W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych: - Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet - godz. 10, - Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Poszukiwaczy - godz. 12, - Parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu - godz. 12, - Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa - godz. 13, - Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - godz. 14. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 6 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Uprzejmie proszę o zadanie pytania panów posłów Waldemara Andzela oraz Marka Polaka z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Odpowiedzi będzie udzielała podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani minister Barbara Socha. Bardzo proszę, panie pośle. Mimo lekkiego wzrostu wskaźnika dzietności nasze społeczeństwo zacznie coraz silniej się starzeć, co będzie oznaczało, iż coraz mniej osób będzie pracowało na emerytury rosnącej liczby osób starszych. Nie brakuje również ostrzeżeń Głównego Urzędu Statystycznego, który napisał o oficjalnym wejściu Polski w okres kolejnego kryzysu demograficznego, który może okazać się o wiele dłuższy niż ten z lat 1997–2007. Dostępne są również szacunki mówiące o tym, że ok. 2060 r. liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie o ok. 60% przy jednoczesnym wzroście liczby osób pobierających świadczenia o praktycznie 100%. Mam pytanie do pani minister: Jakie są przewidziane działania długofalowe mające na celu poprawę bytu polskich rodzin, a co za tym idzie - zwiększenie liczby narodzin, nie biorąc pod uwagę obecnie obowiązujących programów, i czy są już inne projekty, które mają na celu poprawę warunków życia Polaków? Tak, tak. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! W Polsce w 2016 r. urodziło się 13 tys. dzieci więcej niż przed rokiem, a w roku 2017 wzrost urodzeń osiągnął poziom 20 tys. Dostrzegły to hiszpańskie media, które przypisują ten pozytywny trend efektom kilku programów społecznych, zwłaszcza programu 500+, ale wskazują też, że na jedną kobietę w wieku rozrodczym w Polsce przypada 1,4 dziecka, a w Hiszpanii, która ma jeden z najniższych poziomów urodzeń, przypada 1,3. Wynika z tego, że pomimo systematycznego wzrostu urodzeń nadal pozostajemy w kryzysie demograficznym. Dlatego chciałbym zapytać panią minister, jakie dalsze działania zamierza podejmować rząd, aby zażegnać tę nadal niekorzystną sytuację demograficzną. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. O odpowiedź proszę panią minister Barbarę Sochę. Panie Marszałku! Panie Posłanki!

To znaczy, że nasze dzieci, te młodsze, przedszkolne dzisiaj, dożyją tego czasu, kiedy prawdopodobnie w Polsce będzie 21 mln osób.

Starzenie się polskiego społeczeństwa jest faktem i jest to proces bardzo dynamiczny. Według naszych danych już w 2050 r. polska populacja będzie jedną z najstarszych. Zmniejsza się liczba kobiet w wieku rozrodczym. Pomiędzy 2013 r. a 2050 r. liczba kobiet w wieku rozrodczym, czyli od lat 15 do 49 lat, spadnie o 38%.

Tak jak pan poseł wspomniał, współczynnik dzietności od tego najniższego poziomu, z którym mieliśmy do czynienia w 2015 r., kiedy wynosił poniżej 1,3 - który jest uznawany przez demografów za bardzo niski poziom - wzrósł do 1,45, i to jest spora różnica w dobrym kierunku. Oczywiście to jest o wiele, wiele za mało.

Powiem więcej: nawet gdybyśmy przy użyciu czarodziejskiej różdżki zwiększyli dzisiaj dzietność w Polsce dwukrotnie, do takiego poziomu, jaki jest w Izraelu, czyli powyżej trzech, to i tak przez najbliższe lata zmagalibyśmy się z ujemnym przyrostem naturalnym.

To nie oznacza, szanowni państwo, że my będziemy się temu biernie przyglądać.

To prawda. Jest kilka rzeczy, które Platforma Obywatelska zaczęła realizować, chociażby wydłużenie.

Chciałam zauważyć, że podczas kadencji Platformy, przez pierwsze 4 lata działania tego programu powstało 15 tys. miejsc. Środki zwiększono trzykrotnie. To jest oczywiście wszystko za mało. I dlatego, proszę państwa, na początku tej kadencji pan premier Morawiecki zapowiedział przygotowanie wielkiej strategii demograficznej.

Gratuluję. Zapraszam pana posła. Panie Marszałku! Pani Minister! Czy są podejmowane kroki, aby rozbudować infrastrukturę żłobkową oraz ułatwić otrzymywanie dotacji na ich otwarcie? Dziękuję. Pan poseł Marek Polak. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Kraje skandynawskie w przeciwieństwie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie mają problemów z dzietnością i wydaje się, że jest to wynikiem szerokiej dostępności publicznej opieki nad dziećmi poniżej 3. roku życia, a także ułatwiania powrotu na rynek pracy matkom i funkcjonowania elastycznych form zatrudnienia, np. w niepełnym wymiarze czasu, co u nas jest rzadkością. Stąd moje pytanie: Czy zamierzamy korzystać z rozwiązań i wzorców krajów skandynawskich w celu osiągnięcia wyższego wskaźnika urodzeń? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panom posłom. Pani minister - 3 minuty. Zapraszamy.

Są to kraje skandynawskie, ale jest to też Francja, która bardzo, bardzo długo, od wielu dziesięcioleci prowadzi bardzo aktywną i rozbudowaną politykę prorodzinną.

Co do pytania pierwszego, dotyczącego programu rozbudowy sieci żłobków i instytucji, które mają służyć opiece nad małymi dziećmi, oczywiście będziemy te programy rozwijać.

Jak tylko będziemy mogli się podzielić konkretnymi pomysłami, to na pewno państwo posłowie się o tym dowiedzą. Dziękuję serdecznie, pani minister. Dziękuję panom posłom. Tak brzmi regulamin, tak że przykro mi. Proszę państwa, posłowie Jakub Rutnicki i Kazimierz Plocke z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska postanowili zadać pytanie w sprawie podjęcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi natychmiastowych działań, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie całego kraju. W imieniu ministerstwa rolnictwa odpowie sekretarz stanu pan minister Szymon Giżyński. Bardzo proszę pana posła Jakuba Rutnickiego o zadanie pytania. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Jest wielka obawa, ponieważ od czasu gdy wirus ASF pojawił się na terenie województwa lubuskiego, nieopodal Wschowy, w wyniku też opieszałości działań ten wirus się rozprzestrzenia, panie ministrze, sytuacja się nie zmienia. Jestem po rozmowie z samorządowcami, jeszcze z dzisiejszego poranka.

I o to cały czas, panie ministrze, jest wielka prośba.

Tu naprawdę potrzeba wielkich, gigantycznych działań, panie ministrze.

Tak że oczekujemy konkretnych działań. Nie daj Boże, panie ministrze, ale jeżeli ten wirus pojawiłby się w jakimś gospodarstwie, czy państwo zagwarantujecie pomoc finansową i odszkodowanie dla rolników? Oni chcą to od państwa usłyszeć. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Panie ministrze, zapraszam.

Szanowni Panie i Panowie Posłowie! Reakcja była natychmiastowa i wszystko, co się dzieje, dzieje się pozytywnie w formule: natychmiast. Jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie, zagrożenie tam pojawiło się wtórnie w stosunku do województwa lubuskiego.

Ale przecież było wiadomo, że walczymy na terenie obcym, gdzie już pewne rzeczy mogły zajść kilka tygodni temu. Powstał natychmiast płot, ogrodzenie czy przegroda między województwem lubuskim a wielkopolskim, o długości w tej chwili ponad 100 km.

To był jeden przypadek, i tak się natychmiast stało, i drugi przypadek, i też tak się natychmiast stało. To są ogrodzenia doklejone do tej przegrody między województwem lubuskim i województwem wielkopolskim. A więc tam dokonujemy tego samego. Posłużę się przykładem wielokrotnie używanym, ale nie nadużywanym, bo nigdy dość przypominania, że to, co realizowaliśmy i realizujemy w województwie lubuskim i teraz w województwie wielkopolskim, to jest dokładna replika przypadku czeskiego, czyli sposobu, w jaki Czesi poradzili sobie skutecznie z ASF-em - pełna izolacja i likwidacja, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, krok po kroku, tydzień po tygodniu. Inspektorzy Unii Europejskiej na bieżąco to kontrolują, i to kontrolują też skutecznie, nie mają zresztą przesadnych uwag.

Jest to skuteczne, wirus jest osaczony, nie ma w tej chwili żadnych racjonalnych powodów, żeby myśleć, że on się przedostanie.

Mówimy oczywiście o pomocy finansowej. Natomiast na dzisiaj jest tak, że zrobiliśmy literalnie wszystko, zgodnie ze wszystkimi dyrektywami i procedurami, co wykonać należało.

Ale zanim do tego dojdzie w sensie takim, że będziemy mieć już te prawne środki, całkowicie gwarantujące realizację pewnych konkretnych pomysłów, to chcę powiedzieć, że właśnie w kontekście Wielkopolski, w kontekście województw dolnośląskiego, lubuskiego, to co będzie bardzo jasno opisane w ustawie, już praktycznie się dzieje i stanie się. Na mocy decyzji pana premiera, na mocy decyzji ministra infrastruktury grodzimy te przejścia, tak żeby nie było najmniejszej możliwości migracji zakażonych dzików.

Jest to absolutnie pewne zabezpieczenie, żeby wirus się nie rozprzestrzeniał. Bardzo mocno postępują kontrole bioasekuracji.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Po drugie, czy będą zwiększone środki finansowe na działalność Inspekcji Weterynaryjnej w budżecie na rok 2020? Po trzecie, kiedy rząd wprowadzi 100-procentowy zwrot kosztów bioasekuracji w małych gospodarstwach rolnych? Przypomnę, że teraz jest to 50%. Po czwarte, chciałem się spytać, czy rząd planuje uruchomienie ogólnopolskiej akcji informacyjnej skierowanej do konsumentów, do polskiego społeczeństwa w zakresie informowania o skutkach choroby ASF.

Dziękuję. Panie ministrze, zapraszam.

Proszę państwa, Agencja Rozwoju Przemysłu złożyła bardzo korzystną ofertę zakupu przedsiębiorstwa spółki, kontynuacji działalności i rozwiązania podstawowych jej problemów wynikających, jak powiedziałem, z zaszłości historycznych. Jednakże wskutek postanowień sądowych, które blokowały spółce pozyskanie pożyczek, oraz wobec uchylenia uchwały rady wierzycieli te działania restrukturyzacyjne nie mogły być wdrożone. Odpowiadam wprost na pytanie pana posła o przyszłość firmy. Pamiętajmy, że upadłość jest także pewnym narzędziem restrukturyzacyjnym. Naszą intencją jest wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki, kontynuowanie działalności, dlatego że spółka dzisiaj posiada dwa kontrakty, które będzie w stanie realizować. Spółka oczywiście w tym łańcuchu dostaw planowanych dla rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce odegra istotną rolę, jestem o tym głęboko przekonany, więc ma przed sobą przyszłość, ale te zaszłości wymagają oczyszczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Bardzo dziękuję za tę informację.

W związku z tym moje pytanie jest następujące: Czy w tym zakresie były prowadzone jakieś rozmowy z partnerem prywatnym, ażeby zmienić umowę spółki i żebyśmy rzeczywiście mieli możliwość podnoszenia kapitału i być może w inny sposób funkcjonowania?

Wysoki Sejmie! Dziękuję za te pytania, bardzo konkretne, bardzo merytoryczne. Powiem tak: rozmowy z udziałowcem zagranicznym były prowadzone - nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów tych rozmów - ale one nie doprowadziły do konsensusu. Tutaj postawa udziałowca była dosyć zdecydowana i to jest też jedna z przyczyn tej trudnej sytuacji.

Nie zawsze tak jest, że inwestor musi być właścicielem wszystkich podmiotów, które go zaopatrują w procesie konstrukcji farm. Wydaje się, że tutaj nie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją. Powiem tylko, że pracujemy nad takim rozwiązaniem, które pozwoli skupić podmioty Skarbu Państwa w jednym ręku, te podmioty, które będą aktywne w zakresie budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Dziękuję panu ministrowi. Chciałem serdecznie przywitać panów posłów Jana Łopatę.

Cześć, chłopaki i dziewczyny! Witam serdecznie! Proszę, panie pośle. Zapraszam. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Niestety to już ma miejsce. A problem jest ogromny, na razie na etapie składania deklaracji, ale za chwilę będzie trzeba wyciągnąć grosz z portfela, a to są już niestety duże pieniądze i ciągle ich ilość wzrasta.

Związek Gmin Lubelszczyzny, jedna z korporacji, przygotował bardzo dobrą analizę, w której wykazuje się, że do czynników wpływających na wzrost opłat zalicza się cały szereg składowych, m.in. właśnie wzrost stawek za przyjęcie odpadów do instalacji komunalnych, niewystarczające możliwości termicznego przetwarzania odpadów i brak możliwości efektywnego zagospodarowania RDF-u, konieczność dostosowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do zmian legislacyjnych, nieszczelność systemu, brak konkurencji na rynku lub niewystarczająca konkurencja, rosnące ceny energii, transportu, pracy, akcyzy na paliwo, ale również ograniczone - to jest ostatni taki element, zdarzenie na rynku - możliwości zbytu odpadów wyselekcjonowanych.

Otóż postulują oni, by umożliwić rozwój instalacji zgazowywania i utylizację RDF-u, wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (Dzwonek) z tytułu wytwarzania danego produktu, zmniejszenie bieżących obciążeń, oznakowanie produktów i, co podkreślają, edukację. Dziękuję bardzo. Bardzo pięknie pan zdążył, panie pośle. Zapraszamy pana ministra Ireneusza Zyskę. Eh, mógł pan tego nie mówić, panie pośle. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Ministerstwo Środowiska, a obecnie Ministerstwo Klimatu, wdrożyło już szereg rozwiązań, które mają umożliwić gminom bardziej efektywne realizowanie działań w zakresie gospodarki odpadami oraz obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów i w konsekwencji opłat pobieranych od mieszkańców. Zostały one wprowadzone ustawami przyjętymi w lipcu 2019 r., które weszły w życie we wrześniu ubiegłego roku. A zatem efekty ich realizacji będą dopiero widoczne po pełnym wdrożeniu wprowadzonych mechanizmów. Zanim jednak przedstawię państwu posłom te rozwiązania, chciałbym przypomnieć, jakie są przyczyny sytuacji, z jaką mierzą się samorządy w Polsce w zakresie gospodarki odpadami. Do 2012 r. funkcjonował w Polsce system komercyjnych dwustronnych umów pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorcami.

W ramach kosztów przedsiębiorcy określali najczęściej niestety tylko koszty transportu i deponowania odpadów na składowiskach lub, co gorsza, w miejscach nielegalnych, jak np. wyrobiska po żwirowiskach. Dlatego przez wiele lat opłaty dla mieszkańców były niskie w tamtym czasie.

Była to znana nam wszystkim opłata marszałkowska, którą następnie podwyższano kolejnymi uchwałami sejmików samorządów wojewódzkich. To spowodowało, że ceny za odbiór odpadów komunalnych musiały wzrastać. Natomiast niestety muszę ze smutkiem zauważyć, że zmiany wtedy dokonane, w tym jeszcze wcześniej ustawa przyjęta w 2012 r. przez rząd czy większość parlamentarną Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, zlikwidowały w ramach nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. instytucję in-house. To znaczy przedsiębiorstwa komunalne, które do tamtego czasu zajmowały się gospodarką odpadową, odbiorem odpadów, składowaniem odpadów zostały. To spowodowało, że doszło do zmów cenowych, na co wskazują postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doszło do tworzenia takich oligopoli czy nawet monopoli i niestety skutkowało to zmowami cenowymi, które powodowały również wzrost cen za odbiór odpadów komunalnych. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostali objęci wszyscy mieszkańcy, w tym obligatoryjnie właściciele nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców i, fakultatywnie, niezamieszkałych. Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów zaczęły określać rady gminy. Widzę, że czas bardzo szybko płynie, więc chcę powiedzieć, że niestety rząd PO-PSL odroczył wejście w życie tych przepisów związanych z podwyższeniem opłat za korzystanie ze środowiska na bliżej nieokreśloną przyszłość, rok 2015. Dopiero po wyborach rząd Prawa i Sprawiedliwości musiał się zmierzyć z tą tematyką i doprowadzić do wywiązania się z umowy z Komisją Europejską. Natomiast w 2016 r. dokonaliśmy nowelizacji, która spowodowała, że gminy mogły posiłkować się, korzystać z przedsiębiorstw komunalnych w ramach tzw. in-house bez konieczności organizowania przetargów. Ale, proszę państwa, umowy, które po przetargach funkcjonują, były zawarte na 3–4 lata i te skutki w czasie jeszcze trwają. Dopiero kiedy umowy się zakończą, a też będzie dobra wola samorządów, czyli rad gmin, i oczywiście organów wykonawczych gmin: wójtów, burmistrzów, prezydentów, będzie można przystąpić do tego, żeby odbudować ten system in-house.

Dodatkowo w ubiegłym roku, właśnie w roku 2019, dokonaliśmy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach i poprzez zniesienie obowiązku regionalizacji w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych. To bardzo istotna sprawa, ponieważ wcześniej ten mechanizm regionalizacji był bardzo niekorzystny dla samorządów, dla jednostek samorządu terytorialnego. On powodował wymuszenie. Jeżeli dana gmina była skazana na dostarczenie odpadów do konkretnego składowiska (Dzwonek) czy przetwarzania odpadów, to była skazana też na koszty narzucone przez ten podmiot. Super, dzięki bardzo. O pytanie dodatkowe proszę pana posła Mieczysława Kasprzaka. Dziękuję, panie marszałku.

Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Panie ministrze, zapraszam uprzejmie. Dziękuję, panie marszałku. Panie pośle, muszę powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, Ministerstwo Klimatu, a wcześniej Ministerstwo Środowiska, dbają o polskie społeczeństwo, o interes samorządów terytorialnych. Nie chciałbym być uszczypliwy, ale to właśnie polityka poprzedników, której skutki w tej chwili się realizują, doprowadziła do wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych.

To mafia śmieciowa, która dokonała kartelizacji, podziału rynku.

Chcę już dzisiaj zapowiedzieć, że będziemy konsekwentnie bronić tego, żeby te przepisy weszły w życie, bo naszym zadaniem jako Ministerstwa Klimatu jest ochrona interesu społecznego, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Między innymi ustawa z ubiegłego roku, która weszła w życie we wrześniu 2019 r., nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach, daje możliwość zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami przy wykorzystaniu środków finansowych pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych selektywnie. Gminy. No tak.

Z tym jest związany pewien wysiłek, który samorząd terytorialny musi ponieść, ale to jest odpowiedzialność samorządu. Zgodnie z ustawą (Dzwonek) to samorząd terytorialny ponosi odpowiedzialność za gospodarkę odpadami na swoim terenie.

Dziękuję serdecznie.

Przechodzimy. Panie ministrze, powiedzieć jedno zdanie zawsze pan może, bo lubimy się i szanujemy. Mieszkańcy zapłacą mniej za odpady, jeżeli samorządy będą w tym zakresie współpracować z rządem. Dziękuję bardzo. Obowiązek współpracy na pewno leży i na jednych, i na drugich. Tym razem proszę uprzejmie panów posłów Jarosława Gonciarza i Wojciecha Szaramę z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o pytanie w sprawie dofinansowania tzw. systemu deszczowego przeznaczonego do zatrzymywania wód opadowych. Odpowiadał będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu pan minister Ireneusz Zyska, którego już poznaliśmy przy odpowiedzi. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Biorąc pod uwagę zasoby wody, jakimi dysponuje świat oraz nasz kraj i analizując powszechnie dostępne dane, widzimy, że ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca jest u nas poniżej oczekiwań. Coraz powszechniejszym zjawiskiem jest także informowanie mieszkańców, głównie mniejszych gmin, o występowaniu braków wody, szczególnie w okresie letnim. Wiele miast i gmin decyduje się na wdrażanie programów, dzięki którym tworzony jest system deszczowy przeznaczony do zatrzymywania wód opadowych. Ma to na celu ograniczenie nawet o połowę zużycia uzdatnionej wody pobieranej z miejskich wodociągów, odciążenie miejskiej kanalizacji oraz zmniejszenie ryzyka miejskich powodzi i podtopień. Na tego rodzaju niezbędne dziś programy stać przede wszystkim bogatsze gminy. Pragnę jednak zapytać, czy ministerstwo analizowało możliwość uruchomienia swojego programu, którego efekt byłby wymierny. Dziękuję serdecznie. Panie ministrze, zapraszam.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Bardzo dziękuję za to pytanie, niesłychanie istotne z punktu widzenia polityki klimatycznej, związane z gospodarowaniem wodami opadowymi. Jak wiemy, w Polsce niestety z uwagi na zmiany klimatyczne postępuje obniżanie się poziomu wód gruntowych oraz występowanie rok do roku susz w okresach letnich. W odpowiedzi na pytanie chciałbym poinformować, że Ministerstwo Klimatu, a wcześniej Ministerstwo Środowiska, wspólnie z interesariuszami działającymi w obszarze ochrony środowiska, ekologii oraz klimatu prowadzi działania mające na celu zabezpieczenie jednostek samorządu terytorialnego przed negatywnymi skutkami zmian klimatu, w tym przed zmianami dotyczącymi obszaru zrównoważonego i zaadoptowanego do zmian klimatu gospodarowania wodami opadowymi na terenach jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Środowiska opracowało „Politykę ekologiczną państwa 2030” Jest to strategiczny dokument, strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej, która została przyjęta uchwałą Rady Ministrów 16 lipca 2019 r. Polityka ekologiczna państwa jest najważniejszym dokumentem strategicznym w tym obszarze. Jej rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców. Wśród kierunków interwencji polityki ekologicznej państwa znajdują się m.in. adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych. Polityka ekologiczna państwa przewiduje, że działania adaptacyjne będą polegały m.in. na wsparciu opracowania i wdrażania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, budowy niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji. Działania będą również ukierunkowane na zarządzanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych poprzez różne formy retencji, rozwój infrastruktury zieleni, ograniczenie zajmowania gruntów oraz zasklepiania gleby. Konieczność podjęcia działań z zakresu zagospodarowania wód opadowych dodatkowo jest wzmocniona przez prognozy zmian klimatu, które przewidują, że częstotliwość oraz intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych, chodzi zwłaszcza o nawalne deszcze, ulegnie w najbliższych latach zwiększeniu, a ponadto wydłużą się okresy bezopadowe. Konsekwencją nawalnych deszczów są często powodzie miejskie, tzw. powodzie błyskawiczne, oraz podtopienia powodujące straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, z kolei okresy bezopadowe są powodem wystąpienia suszy, niedoborów wody. W tym kontekście działania przystosowawcze są niezbędne.

We wszystkich 44 miastach będących partnerami projektu jako jeden z najważniejszych obszarów wrażliwych na zmiany klimatu wskazano gospodarkę wodną, w tym przede wszystkim obszar gospodarowania wodami opadowymi. Wynika z tego, że jednym z podstawowych działań zwiększających odporność miast oraz przystosowujących miasta do prognozowanych zmian klimatu w zakresie gospodarki wodnej jest budowa oraz rozwijanie zrównoważonych system zagospodarowania wód opadowych. Zadaniem tych systemów będzie ograniczenie skutków oraz zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz zmagazynowanie, tj. retencjonowanie wody opadowej na okres suszy wraz z systemami jej dystrybucji, w szczególności zastosowaniem rozwiązań w zakresie zielonej i błękitno-zielonej infrastruktury. Zrównoważone systemy pozwolą na spowolnienie odpływu wód deszczowych do zbiorników, zatrzymanie, zretencjonowanie oraz wykorzystanie wód opadowych. Szczególnie należy podkreślić ważna rolę błękitno-zielonej infrastruktury, która poza funkcjami zwiększającymi odporność na zmiany klimatu, pełni w miastach szereg innych funkcji, zwiększając komfort życia mieszkańców, np. jako miejsce rekreacji, wypoczynku, jak również funkcje środowiskowo-przyrodnicze - tworzenie klinów napowietrzających, siedlisk dla zwierząt, korytarzy ekologicznych, zwiększenie poziomu różnorodności biologicznej.

Jedną z ważniejszych funkcji takich systemów zrównoważonych jest zatrzymanie, zretencjonowanie oraz wykorzystanie wód opadowych w miejscu ich powstania, w szczególności za pomocą metod naturalnych. Dotychczas w ramach tego typu projektów zostały zakończone trzy konkursy, w wyniku których podpisano umowy o dofinansowanie z beneficjantami, z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich związkami na kwotę blisko 960 mln zł.

Pytanie dodatkowe zada pan poseł Jarosław Gonciarz. Bardzo proszę, panie pośle. To może dopytam tylko: Czy będą wykorzystywane fundusze w ramach wsparcia środków unijnych na te cele? Dziękuję. Wysoka Izbo!

Nie należy ich lekceważyć, bo widzimy rzeczywiście, że z roku na rok te zjawiska pogodowe w postaci długotrwałych susz, a następnie takich nawalnych deszczy, wyładowań atmosferycznych, nagłych zjawisk pogodowych są bardzo dotkliwe dla społeczeństwa i będziemy podejmować wiele takich zrównoważonych działań w ramach polityki klimatycznej, aby obniżyć skutki, również zapobiegając, monitorując, przewidując pewne zjawiska.

Pragnę poinformować ponadto, że Ministerstwo Klimatu przewiduje wsparcie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego działań dotyczących retencjonowania wód opadowych z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury w ramach obecnie przygotowanej nowej edycji mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tzw. mechanizmu norweskiego na lata. Mamy początek roku, ale w tym roku należy się spodziewać przygotowania kompletnej dokumentacji ogłoszenia konkursów, dlatego też apel z tego miejsca do samorządów, jednostek samorządu terytorialnego, aby śledziły prace Ministerstwa Klimatu. Myślę, że w tym zakresie ta nasza współpraca powinna być bardzo spójna, zaawansowana dla dobra obszarów zurbanizowanych, dla dobra mieszkańców miast. Warto również dodać, że możliwość dofinansowania działań z zakresu zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi oraz rozwijania błękitno-zielonej infrastruktury w miastach została zapewniona w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki z możliwością umorzenia. Tak że, panie pośle, szanowni państwo, jestem przekonany, że w tym zakresie, podobnie jak w przypadku gospodarki odpadami, o której mówiłem w poprzednim (Dzwonek) punkcie, dobra współpraca samorządów terytorialnych z rządem przyniesie dobre rezultaty dla dobra mieszkańców. Dziękuję panu ministrowi za wyczerpującą odpowiedź. Dziękuję za przybycie na posiedzenie Sejmu. Teraz posłowie Michał Gramatyka i Marta Golbik z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska zadadzą pytanie w sprawie faktycznego stanu realizacji programu dla Śląska ministrowi funduszy i polityki regionalnej. Zapraszam pana posła, a w międzyczasie witam dzieciaki na galerii. Cześć, dzieci. Zapraszam. Szanowni Państwo! Po 2 latach realizacji tego programu i po kilkunastu tygodniach oczekiwania na informację publiczną udało mi się zdobyć podsumowanie 2 kwartałów 2019 r. Lektura tego protokołu, tego podsumowania, skłania mnie do postawienia następujących pytań: Jaka jest prawdziwa kwota środków, które zainwestowali państwo w województwo śląskie w okresie działania programu? Ale co to znaczy? Bo jeżeli policzymy w kartach poszczególnych projektów środki realnie wydane, to otrzymujemy 8 mld, z czego lwia część to budowa autostrady A1 oraz produkty kredytowe i gwarancje państwowych banków. Jak państwo rozumieją pojęcie środków zaangażowanych? Bo mam wrażenie, że inaczej niż wszyscy. W moim ulubionym np. ze względów semantycznych projekcie inteligentnej kopalni entuzjastycznie raportowane zaangażowanie to 700 mln zł. Realnie wydano niecałe 10. Żaden z 17 podprojektów nie został ukończony, realizację jednego można uznać za zaawansowaną. Wśród ryzyk wykazana została oczywiście kwestia pozyskania finansowania. Jeszcze bardziej niepokoi porzucanie projektów o charakterze innowacyjnym. W myśl państwa protokołu nie będzie instalacji zgazowania węgla, nie będzie instalacji produkcji wodoru, nie będzie instalacji utylizacji gazów pokopalnianych. Odeszliście państwo od tych projektów. Jeszcze bardziej niepokoją zapisy typu: dane utajnione. Finalne pytanie: Dlaczego ten protokół (Dzwonek) nie jest dostępny publicznie? Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana ministra.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

To znaczy to jest program, który cały czas żyje, do którego można dopisywać nowe elementy, o które oczywiście zabiegamy i o które tak naprawdę państwa prosimy. Jeżeli są dobre, to z pewnością będziemy mogli je dodać do programu dla Śląska. A te, które zostały niegdyś wpisane, a okazuje się, że z jakichś powodów nie mogą być zrealizowane, bo np. zmieniła się polityka którejś z firm, które zostały dopisane, z oczywistych względów w tym programie nie powinny się znajdować, ponieważ byłby to program, który nie funkcjonuje. Chodzi o to, żeby w tym programie funkcjonowały tylko te inwestycje, te rozwiązania, które są do zrealizowania.

Po ostatniej aktualizacji w październiku 2019 r., to jest najświeższa informacja, program liczy już 116 przedsięwzięć, których wartość szacowana jest na 62 mld zł. 48 mld zł z tej kwoty to środki, które już pracują w gospodarce. Liczba realizowanych przedsięwzięć, a także skala zaangażowanych środków, czynią z tego programu największe przedsięwzięcie w historii polityki regionalnej w Polsce. Warto również dodać, że program dla Śląska oprócz tego, że cechuje się otwartością, o której powiedziałem na początku, jest programem, który funkcjonuje dlatego, że rząd m.in. negocjuje wysokość oraz warunki wsparcia dla tego programu, np. wsparcia dla regionów poprzemysłowych w ramach unijnego „Just Transition”

Zaangażowanie środków wg celów programu dla Śląska prezentuje się następująco. Warto podkreślić, że mamy możliwość wymienienia kilku celów, dokładnie sześciu. Wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie to jest 11 mld zł. Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu - 0,7 mld zł. Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej - prawie 16 mld zł. Cel piąty, wykorzystanie potencjału województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce - 16,3 mld zł.

Otóż kwota, o której pan poseł wspominał, obejmuje wszystkie umowy, które zostały już zrealizowane w ramach tego programu, ale również te, które są zakontraktowane. Inaczej mówiąc, wliczamy w to również wszystkie inwestycje i działania, które np. w ramach programu „Infrastruktura i środowisko” czy w ramach innych programów zostały zakontraktowane, lub umowy zostały podpisane, a nie są jeszcze rozliczone, co wydaje się dosyć naturalne. To znaczy, że jeżeli wliczamy w to środki, które zostały przeznaczone, i alokacja już występuje, to wpisaliśmy to w ramach kwot, o których mowa, i stąd jest różnica, o której pan poseł powiedział. Dotychczasowe wybrane efekty realizacji naszego programu to jest dofinansowanie 45 projektów w obszarach m.in. energetyki, motoryzacji, medycyny i przemysłu stalowego. 47 tys. osób poniżej 29. roku życia otrzymało wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych. 31 tys. osób powyżej 25. życia zostało przeszkolonych w zakresie korzystania z Internetu.

Dzięki wsparciu z POPC blisko 120 tys. gospodarstw domowych na Śląsku i 530 jednostek publicznych uzyskało dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Jeżeli trzeba, to oczywiście taką listę mogę nawet tutaj panu posłowi wręczyć. Warto zapoznać się również z informacją wydaną w postaci publikatora, o czym pan mówił. Dziękuję serdecznie. Z tego, co pan mówi - to oczywiście niezłośliwe, co powiem, bo nie chcę być w żaden sposób złośliwy - wynika, że już niedługo do swojego okręgu w Zagłębiu będę jeździł krócej niż 6 godzin. To super. Pani poseł, zapraszam serdecznie. Niestety muszę zmartwić zarówno pana marszałka, jak i Ślązaków. Bardzo przepraszam, oczywiście. Nie da się ukryć, że to program, który powstał przed

Kosztował on 120 tys. zł. Uwaga, odwiedza go średnio 270 użytkowników miesięcznie. Nie powiedział pan, gdzie są zaangażowane te środki, a o to chodziło. Ale może przy okazji odniesie się pan minister (Dzwonek) również do kwestii tego świetnego portalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Panie ministrze, uprzejmie zapraszam. Wysoka Izbo! Ale, panie marszałku, z Warszawy do Bielska-Białej pociąg Pendolino jedzie niecałe 3 godziny 20 minut, więc pan marszałek może jeździ innymi drogami.

Jego głównym celem miało być przede wszystkim informowanie o aktualnym postępie prac w każdym z tych przedsięwzięć. Doskonale wiemy również, że w tym portalu jednym z założeń było powstanie mapy, która będzie pokazywała aktualny przebieg tych prac. W tej chwili czekamy na rozliczenie, które ma nam przygotować Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, tego, w jaki sposób te środki zostały wydatkowane. W związku z tym, jeżeli mogę, bardzo proszę o zwracanie się z takimi pytaniami do strefy. Myślę, że tam będzie można takie informacje uzyskać. Te informacje są ogólnie jawnie. Jeżeli byłyby takie problemy, to proszę się do nas zwrócić. My z pewnością będziemy mogli pomóc w uzyskaniu tych informacji. Dziękuję posłom. Proszę uprzejmie posłów: panią Barbarę Dziuk, Annę Gembicką, Grzegorza Wojciechowskiego i Elżbietę Dudę z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o zadanie pytania w sprawie rządowego programu profilaktyki stomatologicznej oraz dostępności świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży. Odpowiadać na pytania będzie przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pani minister Józefa Szczurek-Żelazko. Państwa posłów witam serdecznie i zapraszam do zadawania pytań. Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W wieku 5 lat tylko co piąte dziecko nie ma próchnicy. Warto wiedzieć, że za jej sprawą pojawia się szereg problemów w okresie, kiedy najmłodsi tracą mleczaki na rzecz zębów stałych, oraz rozwijają się inne choroby i powikłania zdrowotne. Głównym powodem takich sytuacji jest zbyt niski poziom profilaktyki stomatologicznej u najmłodszych. Mając to na uwadze, Ministerstwo Zdrowia podjęło szereg działań z zakresu edukacyjno-zdrowotnego przy współpracy z samorządami. Należy podkreślić, że próchnica zębów mlecznych rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie. Niezaleczone ognisko tej choroby potrafi zaatakować mleczaki jeden po drugim, przenosząc się także na wyrzynające się zęby stałe. Tu mam pytanie do pani minister. Co udało się osiągnąć od momentu wprowadzenia od 2018 r. ministerialnego programu profilaktycznego odnośnie do założeń programowych w zakresie celu głównego oraz celu szczegółowego, tzn. zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach publicznych przez wyposażenie szkolnych gabinetów dentystycznych w sprzęt stomatologiczny i niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń? Dziękuję bardzo. Pani minister, zapraszam bardzo, bardzo uprzejmie. Prawda, że jest miło? Wszyscy się uśmiechają do siebie. Proszę bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Rzeczywiście próchnica zębów jest jednym z głównych problemów, jeżeli chodzi o zdrowie jamy ustnej dzieci i młodzieży. Główną przyczyną występowania tego problemu jest w dużej mierze brak systematycznej profilaktyki, brak badań kontrolnych i oczywiście jest to związane z ograniczoną dostępnością do podmiotów, które udzielają świadczeń w tym obszarze. Dlatego też rząd Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w poprzedniej kadencji, mając świadomość tego problemu, podjął konkretne działania, które mają przede wszystkim zwiększyć dostępność do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, jak również zwiększył finansowanie tychże świadczeń. Do całego programu, który jest realizowany obecnie w Polsce, jeżeli chodzi o poprawę dostępności do świadczeń stomatologicznych dzieci i młodzieży, tak jak mówiłam, przygotowywaliśmy się od kilku lat. Już w 2017 r. Sejm podjął ustawę, na podstawie której zostały zakupione m.in. dentobusy, czyli mobilne gabinety stomatologiczne, po jednym dla każdego województwa. Te dentobusy zostały zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i udzielają świadczeń w całej Polsce. Z roku na rok tych świadczeń jest coraz więcej. Jest również realizowany w ramach tych świadczeń szeroki program promocji profilaktyki zdrowia jamy ustnej i stanowi to bardzo ważny element dostępności do świadczeń zdrowotnych. Równocześnie w roku 2018 Sejm podjął kolejną ustawę, na gruncie której zostały przekazane środki dla samorządów, które są organami prowadzącymi szkoły, w ramach których samorządy mogły, jeżeli widziały taką potrzebę, sfinansować zakup sprzętu niezbędnego do utworzenia gabinetów stomatologicznych w szkołach. I był to moment, kiedy samorządy mogły aplikować o te wnioski. Na ten cel na jeden gabinet przeznaczaliśmy 116 tys. Kolejnym etapem, który gwarantuje, jakby scala cały system opieki nad uczniami, jest ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, która została przyjęta przez Sejm w ubiegłym roku, a rozpoczęła swoje działanie od 12 września owego roku. W tej ustawie kompleksowo regulujemy kwestię opieki zdrowotnej nad uczniami, akcentując w dużej mierze profilaktykę i promocję zdrowia, ale również bardzo wyraźnie wskazujemy zasady, na których mają być udzielane świadczenia stomatologiczne. I w tej ustawie stanowimy m.in., że w celu zwiększenia dostępności do świadczeń mogą być one realizowane właśnie w gabinecie szkolnym, który jest wyposażony w odpowiedni sprzęt, funkcjonuje na terenie szkoły i posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również ta dostępność może być zabezpieczona poprzez zawarcie umowy organu prowadzącego szkołę z gabinetem stomatologicznym działającym w otoczeniu szkoły, który posiada również kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, co oznacza, że te świadczenia są w pełni finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Uzupełnieniem tego systemu miały być właśnie te dentobusy, o których mówiłam. W tej chwili już ten system działa. Wiele szkół podpisało umowy albo posiada gabinety stomatologiczne. Szacujemy, że w szkołach jest ponad 700 gabinetów stomatologicznych, które posiadają kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia i udzielają świadczeń zarówno profilaktycznych, jak i kontrolnych i świadczeń naprawczych. Tutaj chcę przypomnieć, że Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył wycenę świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, zwiększając wagę punktową do 1,5. Również jest zagwarantowane finansowanie w 100% świadczeń dla dzieci i młodzieży. Tak że to jest też bardzo istotny element funkcjonowania tych gabinetów. I oczywiście, jeżeli nie ma w otoczeniu szkoły gabinetu, z którym można by było podpisać taką umowę, dotyczy to szczególnie środowisk wiejskich, czasem małych miasteczek, do dyspozycji są dentobusy. Te dentobusy w tej chwili bardzo dobrze spisują się i realizują swoje zadania. W ubiegłym roku ze świadczeń w dentobusach skorzystało ponad 53 tys. dzieci, stanowi to ok. 20% świadczeń stomatologicznych udzielanych dzieciom i młodzieży. To świadczy o tym, jak były one bardzo potrzebne w środowisku i jak są wykorzystywane. Oczywiście te dentobusy mają ustalane harmonogramy pracy na podstawie wniosków konkretnych samorządów lokalnych kierowanych do Narodowego Funduszu Zdrowia, do oddziału wojewódzkiego, który wspólnie z podmiotem, który zawarł umowę na funkcjonowanie dentobusu, ustala harmonogram wyjazdów czy harmonogram pobytu dentobusu.

Dziękuję uprzejmie, pani minister. Szanowna Pani Minister!

Czy są zauważane jakieś korzyści wynikające z tego programu i jakie to są korzyści? Drugie pytanie.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku!

Badania stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży są przeprowadzane co 4 lata, w związku z tym efekty programu będziemy analizować w późniejszym okresie. Natomiast możemy wskazać, jak wzrosła liczba świadczeń finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeszcze raz chciałabym podkreślić, że wszystkie te świadczenia, zarówno profilaktyczne, kontrolne, jak i naprawcze, są finansowane z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządy nie są obciążane żadnymi kosztami funkcjonowania tego programu.

Natomiast co do współpracy z samorządami - rzeczywiście zdarzają się pewne sytuacje, które wymagają naszego wsparcia, i takim wsparciem służymy. Część samorządowców nie do końca ma świadomość, że te świadczenia są w pełni finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, że nie obciąża to budżetu gminy czy powiatu, więc takiej informacji udzielamy. Często zwracają się do nas z prośbą o informację, z kim mogą podpisać taką umowę, ponieważ w otoczeniu nie działa gabinet bądź też działają gabinety, które nie chcą podpisać takiej umowy, więc nasze sugestie są konkretne.

Jeżeli nie ma takiego w otoczeniu szkoły, to też o tym informujemy. Wielu samorządowców z tego korzysta. Informujemy, że właściwy jest kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Następnie dziecko jest informowane, rodzice są informowani, czy jest potrzeba interwencji stomatologa, czy występują jakieś problemy zdrowotne. Rodzic z dzieckiem może się zgłosić w kolejnym dniu, aby uzyskać to świadczenie. Licznie przybyli posłowie z Koalicji Obywatelskiej, pan Rajmund Miller, Mirosława Nykiel, Mirosław Suchoń, Tomasz Kostuś oraz pan Witold Zembaczyński, pragną zadać pytanie w sprawie trudnej sytuacji szpitalnych oddziałów ratunkowych na obszarze całego kraju. Na to pytanie pragnie udzielić odpowiedzi przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan minister Waldemar Kraska. Zapraszam pana posła Rajmunda Millera o zadanie pytania. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Sytuacja całego systemu państwowego ratownictwa medycznego w Polsce jest wysoce niepokojąca. Brak stanowczej reakcji ze strony Ministerstwa Zdrowia może skutkować w najbliższym czasie wystąpieniem kolejnych dramatycznych sytuacji, które dotyczą ludzkiego zdrowia i życia. Pragnę zaznaczyć, że sprawa działalności SOR-ów jest wybitnym przykładem zakłamywania rzeczywistości przez polityków obozu rządzącego na temat dobrej kondycji finansowej i stabilności systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Jedną z przyczyn obecnej sytuacji jest ustanowienie kolejnych restrykcyjnych regulacji, których spełnienie jest obiektywnie bardzo trudne, szczególnie w kontekście trudnej sytuacji kadrowej w zakresie dostępności lekarzy na rynku pracy oraz niedostatecznego finansowania świadczeń, jakie zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dowodem na powyższe stwierdzenie są również słowa pana prezydenta RP Andrzeja Dudy, który stwierdził w grudniu, że warunki w polskich SOR-ach są nieprzyzwoite. Podkreślić należy, że każdy szpitalny oddział ratunkowy jest częścią systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, a więc systemu, który został stworzony w celu skutecznego zabezpieczenia świadczeń ratowniczych na terenie naszego kraju. Co niezwykle ważne, za funkcjonowanie systemu w obszarze danego województwa odpowiedzialni są wojewodowie i to oni w ramach ustawowych kompetencji opracowują wojewódzkie plany działania systemu ratownictwa, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje minister zdrowia. Mając powyższe na względzie zwracam się do pana ministra z prośbą o interwencję w przedmiotowej sprawie, w szczególności proszę o podjęcie działań umożliwiających poprawę funkcjonowania SOR-ów w naszym kraju. Czy ministerstwo dostrzega, że problem braku kadry medycznej, niedofinansowania SOR-ów oraz gigantycznego zadłużenia szpitali powiatowych, chodzi o 14 mld zł, może nieść wyjątkowo niekorzystne skutki dla pacjentów? Czy w ocenie pana ministra może dojść w najbliższym czasie do zamknięć szpitalnych oddziałów ratunkowych w różnych regionach Polski? Dziękuję. Zapraszam, panie ministrze. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Rzeczywiście szpitalne oddziały ratunkowe są jednym z elementów opieki zdrowotnej w naszym kraju. Osobiście uważam, że jednym z ważniejszych, ponieważ trafiają tam pacjenci w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

Dlatego w połowie ubiegłego roku, czyli 27 czerwca 2019 r., Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie w sprawie szpitalnych oddziałów ratunkowych, które zostało opracowane wspólnie w czasie prac zespołu roboczego z przedstawicielami środowiska medycyny ratunkowej, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i pacjentów, ale także personelu medycznego udzielającego świadczeń medycznych w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Dotyczyły one głównie zbyt długiego czasu oczekiwania w SOR-ach na pierwszy kontakt z lekarzem i nadmiernie wydłużonego procesu diagnostycznego w SOR-ach. Pacjent po pierwszym kontakcie z lekarzem zbyt długo oczekiwał na badania dodatkowe, na konsultacje i na decyzję, co do dalszego postępowania w jego przypadku. Chodziło także o nadmierne obciążenie oddziałów ratunkowych pacjentami, którzy nie byli w stanie zagrożenia życia. Dlatego zdecydowaliśmy się na wydanie tego rozporządzenia, aby doprecyzować obowiązki świadczeniodawców, którzy w swoich strukturach posiadają szpitalne oddziały ratunkowe.

System, który wprowadzamy, jest systemem obsługi pacjenta w szpitalnych oddziałach ratunkowych we wszystkich SOR-ach w Polsce. Chcemy, aby na początek ten system zadziałał w największych SOR-ach w naszym kraju. Lekarze pracujący w SOR sygnalizowali nam, że są dodatkowo obciążeni koniecznością poszukiwania miejsc w oddziałach szpitalnych w celu kontynuowania dalszego leczenia.

Jeżeli takich miejsc w danym szpitalu nie ma, pacjent powinien być przetransportowany do innego szpitala przez transport szpitalny, który powinien być zapewniony przez świadczeniodawcę. To wzbudziło troszeczkę niepokoju i kontrowersji w środowisku.

Z danych, jakie otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia i od wojewodów, wynika, że prawie 80% pacjentów zgłaszających się do szpitalnych oddziałów ratunkowych nie jest w stanie wymagającym natychmiastowej pomocy medycznej, czyli stanie zagrożenia życia i zdrowia.

Dziękuję, panie ministrze.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pan minister właśnie odpowiadał na to, na co miał ochotę, niestety, a prosilibyśmy jednak o udzielenie odpowiedzi, panie ministrze, na pytania, które zostały zadane przez mojego szanownego kolegę.

Czy w ocenie ministerstwa może dojść w najbliższym czasie do ich zamykania, czy są takie sygnały? Po drugie, czy ministerstwo dostrzega, a raczej jaki ma pomysł na ten brak kadry medycznej i niedofinansowanie SOR-ów? Bo to powoduje bardzo niekorzystne skutki dla pacjentów. I pytanie: Czy Kancelaria Prezydenta kontaktowała się w tej sprawie, czy ministerstwo może podjęło jakieś działania, żeby ustalić, co pan prezydent, który stwierdził, że te warunki są nieprzyzwoite, miał na myśli i co należy poprawić? Dziękuję bardzo. Panie ministrze, zapraszam serdecznie. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Nie zdążyłem odpowiedzieć. Byłem osobiście w Opolu, spotkałem się ze wszystkimi dyrektorami szpitali opolskich, z dyrektorami SOR-ów, z wojewodą, z marszałkiem.

To samo dotyczy telemedycyny, gdzie wymagany jest dostęp do tomografii komputerowej, ale opis przez lekarza specjalistę może być wykonywany w trybie telemedycyny i może być przekazywany, czyli też de facto w szpitalu fizycznie nie musi być obecny lekarz radiolog.

Mamy też sygnały, że pozostałe szpitale odciążą ten oddział ratunkowy w pracy, więc myślę, że wszystko w Opolu już jest na dobrej drodze, żeby ten oddział ratunkowy mógł dalej funkcjonować. Ja już mówiłem, proszę państwa, o finansowaniu, bo wiemy, że finansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych jest bardzo ważne. W przyszłym roku finansowanie wzrośnie o 128 mln, czyli o 15% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Finanse są bardzo ważne, ale myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy jest to, żeby pacjenci nie kierowali się tylko do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Rozpoczynamy kampanię informacyjną, aby pacjent wiedział, że ma do wyboru nie tylko szpitalny oddział ratunkowy, ale także nocną i świąteczną pomoc lekarską, lekarza rodzinnego.

Dziękuję posłom. Witam serdecznie posłów Jana Warzechę, Zbigniewa Chmielowca, Fryderyka Kapinosa i Marię Kurowską z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, którzy mają zamiar zadać pytanie w sprawie „Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027” i stanu przygotowań do budowy zbiornika wodnego Kąty - Myscowa. Odpowie na to pytanie przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podsekretarz stanu w tym ministerstwie pani minister Anna Moskwa. Proszę uprzejmie pana posła Jana Warzechę o zadanie pytania.

Zapraszam panią minister. Dziękuję serdecznie za to pytanie. Rzeczywiście jest prawdą, że w Polsce mamy małą ilość wody na mieszkańca, i to jest ta zła wiadomość. Natomiast w tym wszystkim jest też dobra wiadomość - ciągle mamy niewykorzystany potencjał w zakresie retencji, czyli zatrzymywania wody, którą mamy. I to jest tak naprawdę główny problem, dużo ważniejszy niż ilość wody, ponieważ z tymi zasobami wody, które mamy, jeżeli będziemy nimi dobrze gospodarować, jesteśmy w stanie dobrze żyć.

To są na chwilę obecną założenia, przejdziemy następnie do opracowywania już szczegółowego programu. Niemniej jednak już teraz prowadzimy działania i konkretne programy związane z retencją. To są różne inwestycje związane z zasobami wodnymi w Polsce, w większości prowadzone przez Wody Polskie.

Pośród tych dużych inwestycji znajduje się też realizacja projektu Kąty - Myscowa, do którego przejdę potem, zbiornik Wielowieś Klasztorna, Niepołomice, odbudowa Zalewu Zemborzyckiego, różne inwestycje związane z przebudową jazów i śluz i innych obiektów wodnych. Jeżeli chodzi o tę część inwestycyjną, to w programie są 94 inwestycje na łączną kwotę ok. 10 mld. Dodatkowo jeszcze mamy 67 propozycji samorządowych, które są w trakcie konsultacji, mniejszych inwestycji, głównie średnich zbiorników retencyjnych. Przeprowadziliśmy taki dobry program pilotażowy z WWF renaturyzacji Białej Tarnowskiej. Ten kierunek renaturyzacji też chcemy kontynuować. Jednocześnie tworzenie retencji na terenach leśnych, zalesienia, zadrzewiania, retencja glebowa, odtworzenie stawów hodowlanych. Został uruchomiony program budowy małych zbiorników i studni. Z naszej strony jest to program bez decyzji wodnoprawnej, na zgłoszenie wodnoprawne, które ułatwia realizację tej mikro- i małej retencji na terenach wiejskich. Jeżeli chodzi o źródła finansowania tego programu, część z tych inwestycji ma już zabezpieczenie w środkach rządowych, w środkach pożyczki Banku Światowego czy też programu operacyjnego PO IiŚ i w kolejnej perspektywie konsekwentnie będziemy te inwestycje też wpisywać w różne źródła finansowania. Niezwykle ważną inwestycją na mapie tego programu jest zbiornik Kąty-Myscowa, rzeczywiście przez lata obiecywany i omawiany bez realizacji. Tutaj kolejna dobra wiadomość.

Szanowni Państwo! Z wielką radością wysłuchałam tej informacji pani minister, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ponieważ sama kiedyś to przeżyłam, wiem, co to jest susza i co to jest powódź, gdy byłam burmistrzem miasta Jasła, które najbardziej cierpi na braku tego zbiornika, jeżeli chodzi o południową Polskę.

Zatem, pani minister, bardzo proszę, aby czuwać nad tą inwestycją, aby ta inwestycja rzeczywiście się rozwijała.

Koledzy mi mówili, że od 50. Od 100 lat są projekty budowy tego zbiornika, czyli Niepodległa już wiedziała, jak ten zbiornik jest potrzebny, a tymczasem tyle czasu zeszło. Myślę, że rząd Zjednoczonej Prawicy dokona tego, na co czekamy już 100 lat. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Chciałam powiedzieć, że dziękuję za ten głos poparcia i obiecujemy współpracę z panią poseł, ale też z pozostałymi osobami, bo zainteresowanych tym projektem nie brakuje, pełną współpracę i realizację zgodnie z harmonogramem. Dziękuję bardzo. Posłowie Andrzej Kryj i Teresa Wargocka z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chcą zadać pytanie w sprawie realizacji przez samorządy przepisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Odpowiadać będzie przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, sekretarz stanu pan minister Andrzej Bittel. Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Posłowie! Szanowny Panie Ministrze! Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej została przyjęta z wielką nadzieją przez wiele milionów Polaków. Dzięki nowym rozwiązaniom przywracane są zlikwidowane połączenia autobusowe do małych miejscowości, co przeciwdziała wykluczeniu komunikacyjnemu. Odtwarzanie zlikwidowanych połączeń odbywa się we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Z niektórych rejonów Polski napływają jednak informacje, że samorządy nie wykazują zainteresowania odtworzeniem połączeń autobusowych. Z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ogłaszane przez wojewodów nabory kończą się często tym, że dziesiątki milionów złotych pozostają niewykorzystane, a samorządy wyjaśniają, że w obecnej sytuacji prawnej nie są w stanie realizować zapisów ustawowych, z drugiej zaś strony mamy do czynienia z opiniami przewoźników, którzy wykazują wolę uruchamiania takich linii i wskazują istnienie potrzeb w tym zakresie. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją dziwną, bo przecież te środki, które są zabezpieczone - w ubiegłym roku było to 300 mln zł, w tym roku jest to 800 mln zł - pomogłyby naprawdę odtworzyć bardzo wiele takich linii. Mam więc pytanie: Dlaczego taka sytuacja ma miejsce i jak przebiega realizacja przez samorządy zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Panie ministrze, zapraszam. Panie i Panowie Posłowie! Jak pan poseł słusznie zauważył, ustawa z 16 maja o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która weszła w życie 18 lipca 2019 r., stanowi podstawę czy jeden z elementów przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Ta ustawa i zawarte w niej przepisy stworzyły podstawę prawną oraz zapewniły środki finansowe na wsparcie dla samorządów na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w skali całego kraju. Środki finansowe zostały rozdysponowane na województwa z przeznaczeniem na dopłaty do deficytowych linii komunikacyjnych, których funkcjonowanie wynika z potrzeb społecznych. Jednostki samorządu terytorialnego, te szczeble, które wymieniał pan poseł, jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego są odpowiedzialne za uruchamianie połączeń komunikacyjnych na obszarach swoich właściwości miejscowych, z uwzględnieniem interesów pasażerów, innymi słowy, swoich mieszkańców. Środki funduszu wspierają samorządy w organizacji transportu autobusowego, a dopłaty stanowią zachętę do podejmowania działań w tym zakresie. Na zwiększeniu oferty przewozowej na uruchomienie połączeń autobusowych skorzystają pasażerowie, przy czym inicjatywa organizacji transportu publicznego na danym terenie leży wyłącznie po stronie władz samorządowych. Pasażerowie oczekują zwiększenia dostępności komunikacji autobusowej, dzięki której możliwa jest większa mobilność społeczna, aktywizująca regiony wykluczone komunikacyjne. Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu trzeba traktować jako inwestycję również w rozwój gospodarczy. Rolą samorządów jest właściwe rozpoznanie realnych potrzeb transportowych lokalnych społeczności i takie zorganizowanie sieci połączeń komunikacyjnych, które przyczyni się do rozwoju ekonomiczno-społecznego obszarów pozostających w ich właściwościach miejscowych. Odpowiedzialne działanie w tym zakresie po stronie samorządów przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych leży w naszym wspólnym interesie, a środki finansowe zapewnione przez rząd dają szansę na lepszą niż dotychczas ofertę przewozową. Pan poseł pytał o kwestie związane z naborami, o kwestie związane z realizacją.

Jest to postęp, choć ten postęp naszym zdaniem, z poziomu Ministerstwa Infrastruktury, mógłby być bardziej widoczny, bardziej intensywny, ale jest. Samorządowcy stopniowo przekonują się do tego przedsięwzięcia.

W roku 2020 przewozy z wykorzystaniem środków funduszu będą realizowane na obszarze 964 gmin.

Mam tutaj całą tabelkę z rozpisaniem na poszczególne województwa, jak wygląda to w sposób zagregowany.

Warto podkreślić, że fundusz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej jest projektem długookresowym - tak też trzeba go traktować - mającym na celu systematyczne uruchamianie regularnych linii autobusowych oraz sprzyjającym tworzeniu wspólnej i funkcjonalnej sieci komunikacyjnej odpowiadającej na bieżące zapotrzebowanie społeczne we współpracy i z główną rolą samorządu terytorialnego (Dzwonek) w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, dziękuję. Proszę bardzo. Panie Ministrze!

Panie Ministrze!

Może dwa zdania o opinii drugiej strony. Proszę, panie ministrze. Oczywiście tym samorządowcom, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie związane z funduszem autobusowym, należą się ogromne podziękowania, bo oni weszli w ten program z taką myślą, że chcą służyć swojej społeczności lokalnej. Drugie ogromne podziękowania należą się z pewnością wojewodom i pracownikom podległym wojewodom za to, że ten program wdrożyli w ekstraordynaryjnym tempie, w bardzo krótkim czasie.

Z tego miejsca zachęcałbym jednak samorządowców, żeby dokonywali analizy swoich potrzeb i potraktowali tworzenie linii komunikacyjnych jako inwestycję w rozwój swojej małej ojczyzny. Dziękuję serdecznie. Dziękuję posłom. Dziękuję panu ministrowi. Proszę państwa, posłowie Andrzej Gawron, Anna Kwiecień i Jerzy Paul z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chcą zadać pytanie w sprawie wdrażania programu Cyber.mil.pl ministrowi obrony narodowej. Odpowiadał będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pan minister Skurkiewicz, z którym zawsze różnimy się w poglądach, ale robimy to w sposób cudowny. Witam pana ministra. Proszę bardzo posłów. Panie Marszałku! Panie Ministrze! W związku z realnymi zagrożeniami i wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa teleinformatycznego Polski Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje program Cyber.mil.pl.

Panie Ministrze, zapraszam. Może wody panu ministrowi? Panie i Panowie Posłowie! Bardzo dziękuję za to pytanie, bo dzisiaj, przypomnę, cyberbezpieczeństwo jest jednym z priorytetów ministra obrony narodowej, stanowi coraz bardziej istotną dziedzinę funkcjonowania współczesnych państw, współczesnych społeczeństw w związku z co rusz to pojawiającymi się zagrożeniami. To jest obszar, który absolutnie musi być i jest rozwijany. Szanowni Państwo! Od 5 lutego 2019 r. Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje kompleksowy program Cyber.mil.pl, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. Program opiera się na czterech strategicznych filarach. Jednym z nich jest właśnie wielopoziomowa oferta edukacyjna w zakresie szeroko pojętego IT oraz cyberbezpieczeństwa. I kilka słów odnośnie do tych działań, które zostały podjęte. Zwiększone zostały limity przyjęć na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej, jak również na Akademii Marynarki Wojennej na kierunkach związanych z bezpieczeństwem informacyjnym.

Chciałbym się właśnie w ten sposób odnieść do limitu, jaki wtedy, w roku 2015, był na tych uczelniach. Szanowni Państwo!

Przez najbliższych 5 lat mury uczelni wojskowych opuści blisko 2000 oficerów w specjalnościach związanych z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem. Szanowni Państwo!

Absolwenci tej szkoły będą przygotowywani do podjęcia studiów wyższych na kierunkach takich jak IT, kryptologia oraz cyberbezpieczeństwo. Szanowni Państwo! Chciałbym zwrócić uwagę, że zgodnie z założeniami do 2025 r. resort obrony narodowej ma mieć do dyspozycji ok. 2000 podporuczników, absolwentów kierunków cyber oraz kryptologia. W ramach łączenia korpusów podoficerów formowane są szkoły podoficerskie informatyki i łączności z siedzibą w Zegrzu i Toruniu. Wojskowa Akademia Techniczna wraz z partnerami zagranicznymi uruchomiła także studia podyplomowe typu MBA w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem. Szanowni Państwo!

Jest to program pilotażowy, który jest dziś realizowany.

Szanowni Państwo! W roku 2020, czyli z końcem sierpnia br., 10 spośród tych placówek oświatowych kończy zaangażowanie w ramach projektu zielonych garnizonów, dwie kolejne - w roku 2021. My w tym roku, po zakończeniu programu w tych 10 placówkach, poddamy ewaluacji realizację tego programu, tak żeby mieć pełną wiedzę na temat tego, jak ten program był realizowany. W resorcie obrony narodowej przeznaczyliśmy 1200 tys. zł na realizację tego programu, ale chcemy iść dalej, szanowni państwo.

Będzie to program, który będzie również kierowany do szkół ponadpodstawowych. Chcemy, żeby w każdym województwie była jedna taka szkoła wyłoniona przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Mamy również zagwarantowane środki finansowe, niebagatelne środki finansowe na realizację tego programu. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Pan minister niech zostanie, to będzie wygodniej. Dziękuję. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

W kwietniu ub.r. podczas np. akademickich mistrzostw świata w programowaniu zespołowym studenci Uniwersytetu Wrocławskiego zdobyli jeden ze złotych medali i tytuł mistrzów Europy w programowaniu oczywiście. Chciałabym dopytać, w jaki sposób ministerstwo planuje pozyskiwanie informatyków do służby w obronie cybernetycznej właśnie z uczelni cywilnych.

Czy tu też jest ukierunkowanie na wykorzystanie osób, które mają w tym względzie pewne przygotowanie? Panie ministrze, proszę. Pani poseł, bardzo dziękuję za to pytanie, bo w istocie zajmujemy się obszarem wojskowym, ale również zachęcamy studentów, którzy studiują dziś na kierunkach cywilnych, do tego, aby mocniej angażowali się w kwestie dotyczące i cyberbezpieczeństwa, i pogłębionej współpracy z polskim wojskiem i Ministerstwem Obrony Narodowej. Pani poseł, w tej chwili na terenie Rzeczypospolitej już kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi uczy się najpierw w klasach mundurowych, bo o tym też muszę wspomnieć.

Dziś we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizujemy program szkolenia wojskowego dla ochotników - i to jest ważna rzecz - pn. „Legia akademicka” Ten program jest uzupełniony o moduł: cyberbezpieczeństwo. Program ten składa się z części teoretycznej, która obejmuje m.in. przedmioty z zakresu wiedzy wojskowej, a także części praktycznej - odbywają się 3-tygodniowe moduły podstawowe prowadzone w formie szkolenia wojskowego.

Do pilotażowego programu w ramach „Legii akademickiej” dołączyło 61 uczelni wyższych; była to edycja z roku 2018. W roku 2019 dołączyły kolejne uczelnie wyższe, jeszcze raz powtórzę, i państwowe, i prywatne.

Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani poseł, dziękuję panu posłowi, dziękuję panu ministrowi. Dzisiaj było miło, panie ministrze. Proszę państwa, kończymy pytania w sprawach bieżących. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 21. porządku dziennego: Informacja bieżąca. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie wzrostu cen energii oraz polityki energetycznej państwa, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana posła Tomasza Piotra Nowaka. Przeczytałem wszystkie te informacje nie tylko dla państwa, ale i dla siebie, żeby się nie pogubić w gmatwaninie przepisów. Panie pośle, mównica jest pana. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiejszy temat tak naprawdę dotyczy politycznej pułapki polskiej energetyki. Węgiel przedstawiany jest przez rząd jako polska racja stanu, choć coraz częściej pochodzi z Rosji. Ponosimy coraz większe koszty takiej polityki. Energia z węgla drożeje z powodu ratowania klimatu planety i rosnących cen uprawnień do emisji CO2.

Ta pułapka energetyczna prowadzi do klinczu decyzyjnego rządu. Powstał co prawda projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, ale jest to polityczna sierota, nie przyjęto go w poprzedniej kadencji.

Dzisiaj w świetle nowych wyzwań transformacyjnych projekt polityki energetycznej już wymaga daleko idących zmian. Polska energetyka w wyniku tej decyzyjnej niemocy jest niekonkurencyjna.

Stąd coraz większy import energii, przewyższający eksport. Dla gospodarstw domowych, dzięki URE zatwierdzającemu koszty uzasadnione, mamy ceny energii niższe niż u sąsiadów, ale po 2021 r. Polska będzie zobowiązana do uwolnienia cen. Aby nie było to szokujące dla gospodarstw domowych, produkcja energii musi być tańsza dzięki konkurencyjnemu rynkowi, a pomoc publiczna powinna polegać nie na zamrażaniu cen, lecz na stawianiu na tańszą energię.

A ceny energii węglowej będą rosły. Polska staje się więc coraz mniej konkurencyjnym energetycznym skansenem Europy.

Ówczesny prezes URE złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Rodzi to pytanie o to, czy podwyżka cen i ich zamrożenie ustawą w 2018 r. zostały spowodowane tylko zwyżką cen uprawnień i kosztami wydobycia. Jednocześnie spółki obrotu podniosły zdecydowanie opłatę handlową, a od października do rachunku dojdzie 10 zł za miesiąc, jeśli chodzi o koszt opłaty mocowej.

Stąd zdecydowanie trzeba uzyskać społeczne poparcie dla programu sprawiedliwej transformacji energetycznej, ze wskazaniem roku 2050 jako roku gospodarki zeroemisyjnej. Tego wymagają i nasz klimat, i nasze zdrowie, i nasze portfele. Żeby to przeprowadzić, rząd musi po prostu przystąpić do programu sprawiedliwej transformacji energetycznej, a tego niestety nie robi. Żeby sięgnąć po pieniądze, 100 mld euro, trzeba zdecydowanie powiedzieć: tak, chcemy wziąć te pieniądze i chcemy je przeznaczyć na transformację energetyczną. Musimy wyjść z tej energetycznej pułapki, na początek przez kilka zdecydowanych ruchów. Dla regionów górniczych, np. Wielkopolski wschodniej, przygotować rządowy program kompensacyjny. Odblokować energetykę wiatrową na lądzie, pozostawiając władztwo samorządom. Małe i średnie firmy powinny mieć możliwość produkcji energii na własne potrzeby oraz ułatwioną procedurę sprzedaży i zakupu energii w formule bezpośredniej w przypadku odbiorcy końcowego. Rozważyć trzeba wreszcie wprowadzenie dodatkowych taryf czasu rzeczywistego, które umożliwiłyby (Dzwonek) elastyczne zarządzanie podażą i popytem w silnie zmieniających się warunkach. Panie pośle, jakbym miał zadać to pytanie, lepiej bym tego nie potrafił zrobić. A teraz posłuchamy podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pana ministra Tadeusza Skobla. Zapraszam serdecznie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za ten wniosek Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, ponieważ daje to możliwość poinformowania Wysokiej Izby oraz obywateli o programie przeciwdziałania wzrostowi cen energii elektrycznej, który udało się nam wprowadzić i zrealizować w 2019 r., oraz o zarysach mechanizmu na rok 2020, nad którym obecnie pracujemy. Z tego powodu moją wypowiedź podzielę na trzy części. Druga będzie dotyczyła planów rekompensat za wzrost cen w 2020 r. A trzecia będzie dotyczyła polityki energetycznej Polski, o której również usłyszeliśmy we wniosku.

Były również informacje o podwyżkach 68-procentowych.

Samorządy, małe i średnie przedsiębiorstwa, rolnicy, szpitale, stowarzyszenia, odbiorcy cennikowi indywidualni nie zapłacili wyższych cen niż w 2018 r.

Tam, gdzie nie było możliwe zamrożenie cen energii elektrycznej w II półroczu 2019 r. ze względu na ustalenia z Komisją Europejską, zaproponowaliśmy dopłaty w ramach dozwolonej pomocy de minimis. Chodzi tu o średnie i duże przedsiębiorstwa. W 2019 r. żaden odbiorca końcowy energii elektrycznej nie pozostał bez pomocy państwa. Efekt naszych działań widać po danych publikowanych przez Komisję Europejską, dotyczących zmian cen energii elektrycznej między rokiem 2019 a rokiem 2018, które teraz przytoczę. Wzrost rachunków odbiorców indywidualnych powyżej 10% nastąpił w sześciu państwach Unii Europejskiej. Wzrost rachunków powyżej 5% - w 13 państwach Unii Europejskiej.

Dzięki temu mamy jedne z najniższych cen w Unii Europejskiej. To nie jest tylko zasługa rządu Rzeczypospolitej Polskiej, lecz również całego parlamentu, który zebrał się na dedykowanym posiedzeniu 28 grudnia 2018 r. Za ustawą zagłosowało ponad 95% głosujących posłów, a przeciw ustawie głosowało jedynie trzech posłów. Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla parlamentu. Często państwo pytacie również, czy sprawnie realizowane są wypłaty dla spółek obrotu przez Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Przedsiębiorstwa obrotu realizujące obowiązek stabilizacji poziomu cen energii elektrycznej mogą występować z wnioskami do końca stycznia roku 2020, a średnie i duże przedsiębiorstwa mogą występować o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis do końca czerwca roku 2020. Warto w tym miejscu wskazać na sukces prowadzonego dofinansowania w ramach pomocy de minimis dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Pamiętam, jak w czerwcu ub.r. przy okazji nowelizacji posłowie opozycji wątpili w to, że średnie i duże przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie w II półroczu roku ubiegłego. Podmioty te mogą składać odpowiednie wnioski od października 2019 r.

Mechanizm na rok 2020.

Otóż w roku 2018 doszło do zdestabilizowania sytuacji cen na giełdzie energii elektrycznej, na której nastąpił gwałtowny wzrost cen. Był to efekt głównie skokowego wzrostu cen uprawnień CO2.

Dziękuję bardzo. Do zadania pytań zgłosili się posłowie i posłanki: Ewa Malik, Krzysztof Gadowski, Marek Dyduch, Barbara Dziuk, Aleksander Miszalski, Grzegorz Wojciechowski, Urszula Zielińska, Anna Kwiecień, Gabriela Lenartowicz, Marek Polak, Ewa Kołodziej, Michał Szczerba, Cezary Grabarczyk, Paulina Hennig-Kloska i Paweł Poncyljusz. Czy ktoś z państwa posłów jeszcze chciałby zapisać się do głosu? Czy jeszcze ktoś? Proszę bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Mamy 17 posłów zgłoszonych do zadawania pytań, w związku z czym ustalam limit 2-minutowy. Zapraszam serdecznie.

Pan poseł Krzysztof Gadowski, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja bym chciał zatrzymać się na chwilę przy tej destabilizacji, o której pan mówił, cenowej energii na Towarowej Giełdzie Energii.

W wyniku tego postępowania oczywiście pojawił się wniosek do prokuratury. W międzyczasie w Sejmie, 28 grudnia tego roku, pojawił się projekt ustawy, bardzo słaby, poprawiany później wielokrotnie, który namieszał trochę u przedsiębiorców, u tych, którzy również tę energię sprzedawali.

Chciałbym pana spytać jednoznacznie: Czy znamy już wyniki tego postępowania?

I kiedy to śledztwo zostanie zakończone? Dziękuję serdecznie panu posłowi. Pan poseł Marek Dyduch, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

Mam tego typu pytania: Czy importujemy energię? Jaka to jest wielkość? Czy to wynika z tego, że nasze zasoby są za małe, czy to po prostu jest normalne na rynku europejskim, że część energii się kupuje? Po drugie, jeżeli chodzi o inwestycje,

To są ogromne nakłady, Niemcy poważnie to traktują, w każdym landzie jest departament, który zajmuje się właśnie energią cieplną. Czy my w tę formę energii odnawialnej będziemy inwestować?

To jest ważna informacja też w kontekście naszych planów inwestycyjnych. Chciałem jeszcze dopytać o jedną rzecz: Czy te nowe bloki energetyczne w Opolu i w Jaworznie to są odnawiane bloki, które były, czy są to wybudowane nowe bloki w ramach istniejących już elektrowni? Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Proszę pana posła Jana Łopatę z klubu parlamentarnego PSL-Kukiz15. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W poprzednim punkcie obrad Sejmu w tzw. pytaniach w sprawach bieżących pytaliśmy z kolegą o bardzo ważny społecznie element życia, a mianowicie o ceny wywozu odpadów, segregacji odpadów.

Więc pytanie, które się ciśnie: Czy samorządowcy w roku 2020 mogą liczyć, przynajmniej w tym zakresie firm segregujących, na jakieś rekompensaty za wzrost cen energii?

A oczywiście z przyczyn regulaminowych, o których wcześniej rozmawialiśmy, nie mógł pan przedstawić polityki energetycznej państwa, bo wydaje się, że tu jest może i ważniejszy element.

Bo to, że my importujemy energię, to jest wiadomo, ale przecież w Polsce są zasoby, źródła energetyczne i warto to wykorzystać, wydaje się, sprzedawać, a nie importować. Dziękuję panu marszałkowi za udzielenie głosu. Dziękuję panu posłowi za miłe pytanie. Bardzo proszę. To już nie pierwsze pytanie pani poseł, dzisiaj. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Polityka energetyczna przyjęta obecnie przez rząd z ramienia Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim jest ukierunkowana na bezpieczeństwo energetyczne i kogenerację energetyczną. W związku z tym mam do pana ministra pytanie z zakresu energetyki odnawialnej, która też jest, bym powiedziała, jednym z głównych kierunków rozwojowych w Polsce. Ta właśnie energetyka odnawialna musi następować w sposób ewolucyjny z zagwarantowaniem źródeł rezerwowych zależnych od warunków pogodowych. Gaz jest jednym z tych surowców mniej emisyjnych, które mają zapewnić ewolucyjną transformację. Jest jednocześnie paliwem pochodzącym głównie z importu. Czy realizowane inwestycje gazowe pozwolą na pokrycie wzrastającego zapotrzebowania na gaz w elektroenergetyce i ciepłownictwie? Jaka jest zależność energetyczna Polski?

Mam pytanie dotyczące odbiorców indywidualnych, dla których ceny energii nie są zatwierdzane przez prezesa URE. Na przykład korzystający z prawa do zmiany sprzedawcy i cen rynkowych objęci będą mechanizmem kompensowania podwyżek. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! To, że ceny energii będą w Polsce rosnąć, było wiadomo długo przed waszym dojściem do władzy i rząd Platformy i PSL-u chciał Polskę na ten fakt przygotowywać, inwestując m.in. w energię wiatrową, co skutecznie jedną ustawą zaoraliście. Ceny energii na rynku hurtowym w Polsce są najwyższe spośród uprzemysłowionych krajów sąsiednich i od początku tzw. dobrej zmiany te ceny energii w Polsce są średnio o 20% wyższe niż w Niemczech, a dla przedsiębiorstw produkcyjnych cena energii to jeden z głównych, kluczowych kosztów działalności. Wzrost cen energii o kilkadziesiąt procent, który może nas wkrótce dotknąć, będzie skutkowało przerzuceniem tego kosztu albo na konsumentów albo ograniczeniem produkcji i w konsekwencji zapaścią gospodarki. W jednym z wywiadów pani minister Emilewicz stwierdziła: przeciętny konsument indywidualny przyjmie znaczącą podwyżkę z niezadowoleniem, ale nie zachwieje ona jego budżetem, natomiast przedsiębiorstwa, takie jak stalownie, najzwyczajniej analogicznej podwyżki nie wytrzymają. W 2019 r. wprowadziliście wprawdzie mechanizm utrzymania cen, ale jak długo można ten problem zamiatać pod dywan. Nie uciekniecie od tego i prędzej czy później wszyscy będziemy musieli tę żabę zjeść, a na końcu zapłacą za to obywatele. Zresztą w Krakowie już płacimy za to, zwłaszcza pracownicy huty ArcelorMittal, ale również Kraków podatkowo. Na moją interpelację w sprawie huty minister Emilewicz odpowiedziała wprost: Przypadek wstrzymania produkcji w oddziale ArcelorMittal w Krakowie jest odzwierciedleniem trudnej sytuacji przemysłu hutniczego w Polsce. Przyczyniły się do tego m.in. wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2. A ja chciałbym zapytać: Ile wynosi koszt rekompensat za wzrost cen energii dla wszystkich przedsiębiorstw w roku 2019?

Dziękuję, panie pośle. Proszę pana posła Andrzeja Szejnę z klubu parlamentarnego Lewica. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Czy zna pan raport 11 tys. naukowców, który ukazał się w magazynie naukowym „BioScience”, który podpisało 11 tys. naukowców ze 153 krajów, który przewiduje ogromne cierpienie ludzkości związane ze zmianami klimatycznymi? Te zmiany klimatyczne oczywiście odnoszą się również do polityki energetycznej, do zasobów naturalnych, do zwiększenia populacji światowej. Odnoszą się również do energii odnawialnej. Chcę panu ministrowi powiedzieć, że nie widzę w polityce rządu jakiejkolwiek refleksji dotyczącej zmian w polityce globalnej, w polityce Unii Europejskiej, nowego paktu zielonego dla Europy. Czy pan minister przewiduje korektę polityki rządu? Pan wie, że kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie umiera pośrednio czy bezpośrednio ze względu na zanieczyszczenie środowiska? Może - zwracam się tutaj do koleżanek i kolegów z klubu Prawa i Sprawiedliwości - jednak dojdzie do was to, że zmiany klimatyczne już nas otaczają i nas dotyczą. Panie ministrze, w ramach zagadnień dotyczących polityki energetycznej: Czy już pan przewidział w budżecie na najbliższe lata, w budżecie rządu - bo będziecie rządzić przez najbliższe lata - środki finansowe na kary, jakie będzie nakładała Unia Europejska na Polskę za to, że nie będziemy wypełniać wymogów i zobowiązań wynikających z udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym Polski?

Moje pytanie do pana ministra jest takie.

Oba te programy powinny być implementowane do polityki energetycznej państwa 2040 r. Brałem udział w opiniowaniu tego dokumentu. Pytanie podstawowe brzmi: Kiedy ostatecznie rząd przedstawi projekt polityki energetycznej państwa? Uważam, że ten, który jest, skrojony jest na miarę państwa polskiego i potrzeb ekologicznych. Natomiast tutaj mam takie dane. Elektrownie cieplne produkują 19 tys., wodne - 300, elektrownie wiatrowe - 3 tys. MW. Jaką mamy sytuację w całym systemie?

Dziękuję serdecznie panu posłowi. Proszę państwa, witam panią marszałek Gosiewską. Ja państwu za dzisiejsze 3 godziny serdecznie dziękuję. Mamy fantastyczne posłanki i fantastycznych posłów. Przepraszam, fotel. Dziękuję, panie marszałku, jak zwykle uroczy. Zapraszam pana posła Grzegorza Wojciechowskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rząd zadeklarował wsparcie dla energetyki rozproszonej i prosumenckiej. Jest to bardzo ważna rzecz, dlatego że energia będzie wykorzystywana w sposób moim zdaniem najbardziej racjonalny, czyli tam, gdzie jest zapotrzebowanie na tę energię, ona będzie produkowana. Koszty przesyłu wyraźnie się zmniejszą.

Na przykład z raportu Schroedera wynika, że w przypadku energetyki wiatrowej ten bilans jest ujemny. Stąd moje pytanie, panie ministrze.

Czy rząd będzie w stanie zapewnić zrekompensowanie podwyżek cen prądu w gospodarstwach domowych w bieżącym roku? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Urszula Zielińska, Koalicja Obywatelska. Zapraszam serdecznie. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni Goście! Szanowni Państwo! 1 stycznia br. upłynęły terminy przesłania przez rząd do Komisji Europejskiej dwóch planów, dwóch ważnych, strategicznych planów: „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”, tzw. strategii krótkoterminowej, i „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2050”, tzw. strategii długoterminowej, wymaganych rozporządzeniem unijnym z 2018 r. Chcę w związku z tym zadać kilka pytań. Po pierwsze, odnośnie do strategii krótkoterminowej. Czy konsultacje publiczne, które państwo przeprowadziliście w terminie od 14 stycznia do 18 lutego, czyli przez 4 tygodnie, spełniły wymagania rozporządzenia dotyczące jakości konsultacji publicznych? Zacytuję: Państwo członkowskie zapewnia wielopoziomowy dialog, w którym aktywnie uczestniczyć oraz - uwaga - dokonywać przeglądu postępów mogą samorządy lokalne, organizacje społeczne itd., itd. Drugie pytanie. Dlaczego w tym planie nie uwzględniliście zaleceń Unii Europejskiej z czerwca zeszłego roku odnośnie do zwiększenia naszej ambicji co do udziału OZE, energii odnawialnej, do 25% na rok 2030? Pytanie: Dlaczego? Czy strategia długoterminowa została przygotowana i przekazana do Komisji Europejskiej w wymaganym terminie, do 1 stycznia 2020 r. O ile mi wiadomo - nie, ale jestem ciekawa, może tego nie znalazłam. Ostatnie pytanie, odnośnie do aktywów państwowych.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Zapraszam. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jestem mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego, jego zachodniej części.

Kopalnie węgla brunatnego są umiejscowione po stronie Wielkopolski, w województwie wielkopolskim, i tam rzeczywiście gminy korzystają ze wszystkich dobrodziejstw związanych z istnieniem tych kopalni, natomiast skutki zauważamy w województwie kujawsko-pomorskim, zwłaszcza te negatywne, przede wszystkim te negatywne, bo pozytywnych tutaj nie ma, a zwłaszcza tych finansowych. Dlatego oczekuję odpowiedzi i informacji, czy rząd zastanawia się nad rekompensatą dla gmin - nie tylko tych gmin, na terenie których są położone odkrywki węgla brunatnego, ale także tych gmin, które znajdują się na brzegu oddziaływania leja depresyjnego. Jest to bardzo ważna kwestia, szczególnie dla rolnictwa, ale także dla funkcjonowania czy turystyki, czy generalnie obszarów leśnych w tamtym rejonie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Opracowana przez rząd polityka energetyczna zakłada intensywny rozwój źródeł odnawialnych, które już w 2030 r. mają dostarczać przeszło 30% energii elektrycznej generowanej w kraju z tzw. OZE. Mają to być w większości turbiny wiatrowe na lądzie i morzu oraz źródła fotowoltaiczne, a więc jednostki uzależnione od bieżących warunków atmosferycznych. Czy w takiej sytuacji zapewnione zostanie bezpieczeństwo dostaw energii do wszystkich odbiorców zgodnie z ich zapotrzebowaniem? Jaki nastąpił przyrost mocy OZE w elektroenergetyce w ostatnich latach w porównaniu do krajów europejskich? Mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ bardzo często pada tutaj z mównicy zdanie odnoszące się do wzrostu cen uprawnień, certyfikatów CO2.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani poseł Gabriela Lenartowicz, Koalicja Obywatelska, z kolejnymi pytaniami. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

W budżecie takiej kwoty nie ma. Rozumiem, że i tak my, odbiorcy końcowi energii elektrycznej, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio, za to zapłacimy. Chciałabym wiedzieć, co rząd przewiduje, z jakich środków to pokryje i w jaki sposób obciąży nas tymi kosztami. A koszty są spowodowane polityką, którą prowadzi rząd PiS. Od 2016 r. praktycznie zablokowano najtańszą energetykę lądową i wiatrową.

To jest obecnie najtańsza na rynku hurtowym energia.

Ten import byłby znacznie większy, gdyby infrastruktura na to pozwalała.

Dziękuję bardzo, pani poseł.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jestem posłem z województwa podlaskiego, gdzie mamy skupione najbardziej rozwinięte rolnictwo, mleczarstwo. Największe zakłady to Grajewo, Piątnica, Wysokie Mazowieckie i wszyscy rolnicy z niepokojem obserwują to, co się dzieje w Ostrołęce. Z jednej strony słyszymy, że zgodnie z planem przebiega budowa elektrowni, bloku C w Ostrołęce, natomiast z drugiej strony zastanawiają się rolnicy, jak to wpłynie na szeroko pojęte rolnictwo.

Są okresy, kiedy rolnicy nie mogą tego wywieźć, natomiast osad pofermentacyjny z biogazowni można przez cały rok wywozić na pole. A funduje nam się za granicą województwa podlaskiego, już na obszarze województwa mazowieckiego, ogromną elektrownię, ogromny blok, gdzie 280 wagonów węgla na dobę będzie przywożonych.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam, panie pośle. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Jak wszyscy wiemy, od czerwca 2018 r. do końca roku 2019 ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie uległy zmianie i były jednymi z najniższych w Europie. Tylko pięć państw wyprzedziło nas w tym rankingu. W tym samym czasie ceny energii w europejskich państwach systematycznie rosły, co jest skutkiem polityki klimatycznej, a także rosnących cen paliw. I myślę, że podobnie może być też w Polsce, bo my również musimy ponosić koszty uprawnień do emisji CO2.

Wysoka Izbo! Wszyscy chcielibyśmy oddychać czystym powietrzem i żyć jak najdłużej. Wszyscy również chcielibyśmy płacić niskie rachunki za prąd. Dlatego rząd bezwzględnie musi zauważyć potrzebę inwestowania w OZE, w tym w przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne. I będę chciała się właśnie na tym zagadnieniu skupić. Bardzo boli mnie to, że rządzący nie traktują poważnie prosumentów. Polityka rządu jest bardzo brutalna, ponieważ pozwala się tylko na inwestycje w mikroinstalacje przydomowe do 10 kW peak, a przy korzystaniu z takiej instalacji nie można zarabiać, tym bardziej że płaci się spółkom energetycznym spory haracz. Przy 10 kW peak to jest 25% energii, którą trzeba oddać spółkom energetycznym, przy większych aż 40% wyprodukowanej energii trzeba oddać. Jest to absolutnie niepodmiotowe traktowanie prosumentów, przedsiębiorczych Polaków.

Dodatkowo bardzo dużym kosztem jest na początku sama inwestycja.

Dlatego mam konkretne pytania: Kiedy rząd planuje znowelizować ustawę o odnawialnych źródłach energii? Czy rząd wreszcie zaufa przedsiębiorczym obywatelom, by mogli bez ograniczeń w ilości kilowatów - mam tu na myśli kilowaty - budować te instalacje? I czy ten współczynnik będzie 1:1, tak żeby traktować prosumenta po partnersku, żeby on nie musiał płacić haraczu spółkom węglowym?

Dziękuję, pani poseł. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Podwyżki cen prądu dla indywidualnych odbiorców nie będzie. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Czyny a słowa. Słowa, które nic nie znaczą, ponieważ fakty są następujące. Wysoka Izbo! W Polsce jest ok. 15 mln gospodarstw domowych, które są odbiorcami energii. Z taryf zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki korzysta prawie 10 mln. No i cóż? Nowy rok - nowe informacje z Urzędu Regulacji Energetyki. Kolejne podwyżki cen prądu stają się faktem. Mówiłem o 15 mln gospodarstw domowych, ale chciałbym, Wysoka Izbo, zwrócić uwagę na gospodarstwa domowe, które tworzą lub współtworzą seniorzy. 35% gospodarstw domowych stanowią właśnie gospodarstwa z udziałem seniorów. I tu sytuacja wygląda katastrofalnie, bo opłaty za mieszkanie, opłaty za prąd stanowią znaczną część dochodów tych gospodarstw domowych. Sytuacja skrajnie się pogarsza wtedy, kiedy mamy do czynienia z seniorami żyjącymi samotnie.

Szanowni państwo, w zeszłym roku było 227 tys. osób, które otrzymywały emerytury niższe od minimalnych gwarantowanych przez państwo. Jak ta sytuacja - i to jest pytanie do rządu - wpłynie na gospodarstwa domowe (Dzwonek), które tworzą seniorzy, których emerytury są poniżej minimalnych gwarantowanych? Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Region łódzki to ważny region na energetycznej mapie Polski. W regionie tym położony jest Bełchatów i znajduje się wielki kompleks wydobywczy, ale także wytwórczy energii elektrycznej. Trzeba powiedzieć, że prądu będzie już niedługo mniej, bo dziś Bełchatów zaspokaja 20% potrzeb energetycznych kraju. Warto dodać, że to jest najtańszy prąd wytwarzany w Polsce. Za 15 lat przestanie być wydobywany węgiel w Szczercowie. W tym zagłębiu i w elektrowni bezpośrednio pracuje dziś 12 tys. pracowników. Co z perspektywą dla Złoczewa? Już dzisiaj trzeba odpowiedzieć mieszkańcom regionu na to pytanie, bo za 15 lat ten region stanie przed perspektywą utraty kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. Na początku dekady lat 90. minionego wieku taka zapaść w branży włókienniczej spowodowała gigantyczny kryzys w stolicy regionu łódzkiego. Jaka perspektywa czeka Bełchatów? Czy jest przygotowywana (Dzwonek) alternatywa w postaci energetyki jądrowej i czy będzie lokalizowana w okręgu bełchatowskim? Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Paulina Hennig-Kloska, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Brak polityki energetycznej kraju i brak transformacji energetycznej tak naprawdę dzisiaj powodują, że musimy płacić coraz więcej za prawa do emisji. Rozumiem, że rząd w zasadzie jest zadowolony, bo przecież te pieniądze z praw do emisji wpływają do budżetu i możecie go skleić. Ale przecież z drugiej strony ktoś to płaci, płacą to tak naprawdę obywatele w cenach towarów kupowanych w sklepie i w cenach rachunków za prąd.

Wraz z brakiem polityki energetycznej kraju i brakiem transformacji energetycznej coraz więcej prądu kupujemy z zagranicy. Energia kupowana z zagranicy pokrywa już 6% zapotrzebowania naszego kraju, i ten udział będzie rósł, nie mamy co do tego wątpliwości. Pod koniec roku zagraniczne elektrownie pokrywały nawet 19% zapotrzebowania Polski na moc. Gdzie ta suwerenność, o którą rząd Prawa i Sprawiedliwości niby cały czas tak walczy?

Dobrze wiemy, że większy import krótkookresowo (Dzwonek) może dać tańszy prąd, ale uzależnianie się od importu to tak naprawdę większa podatność naszego kraju na wzrost cen. Co rząd zamierza z tym zrobić? Panie Ministrze! Zwracam się do pana jako do przedstawiciela rządu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości to rząd, który nie dba o obywateli i konsumentów, jeśli chodzi o ceny energii. Ceny energii rosną, dlatego że zaklinaliście kult węgla i popieracie kult węgla w miksie energetycznym Polski.

To przedsiębiorcy przestają być tak konkurencyjni, jak byli dotąd. To przedsiębiorcy, mając nowe ceny energii, będą musieli oszczędzać. Na kim? Na pracownikach, na swoich rodzinach, na warunkach pracy, na urządzeniach, które będą w tych przedsiębiorstwach. Nie dbacie również o przedsiębiorstwa energochłonne, które niby miały dostawać różnego rodzaju wsparcie, ale symbolem rządów Prawa i Sprawiedliwości w duchu reindustrializacji polskiego przemysłu jest wygaszanie pieca w Nowej Hucie, w Mittalu. Nie dbacie również o państwowe spółki energetyczne.

Nie są w stanie wykonać planów inwestycyjnych, bo nie mają na to pieniędzy. Nie dbacie również o zdrowie Polaków, bo przecież smog generuje cały szereg różnego rodzaju chorób, o czym już wcześniej była mowa. Sami nie wiecie, czego chcecie. Nie dość tego.

A gdzie jest to dla nas? Jest tylko po cichaczu przesłane (Dzwonek) do Komisji Europejskiej. W związku z tym zwracam się do pana z dwoma pytaniami i prośbami. Ukrywacie to przed Polakami?

A więc trochę mniej węgla i ta energia może nie drożeć tak szybko, jak drożeje dziś.

Pani poseł, przepraszam. Pani poseł również. Panie pośle, bardzo proszę. Wysoka Izbo! Tauron podnosi ceny energii o 12%, tzn. że mieszkańcy Bielsko-Białej, Cieszyna, Pszczyny, Żywca i powiatów zapłacą 12% więcej za prąd. Ale to nie wszystko, ponieważ to wpłynie na ceny innych produktów, usług, czyli w sklepach zapłacą więcej za podstawowe artykuły, takie jak chleb, jajka, masło itd.

Bardzo bym prosił o tę odpowiedź. Drugie pytanie dotyczy spółek obrotu energią, tych mniejszych spółek, które funkcjonują, w zasadzie funkcjonowały do pewnego momentu na rynku handlu energią, przyczyniając się do większej konkurencyjności na tym rynku. Zawirowania, które zostały spowodowane przez nieprzewidywalną politykę rządu w tym zakresie, spowodowały, że spółki znalazły się w kłopotach. I teraz pytanie, czy rząd ma jakikolwiek plan na to, żeby te spółki mogły nadal funkcjonować, żeby ten ważny element rynku energetycznego, który można określić jako tworzenie warunków konkurencyjności, jako dostarczanie prądu w w atrakcyjniejszych cenach dla odbiorców, jednak na rynku pozostał, a te spółki nie ogłaszały upadłości, nie znikały z rynku. Bo niestety dzisiaj wygląda to w ten sposób, że działania rządu Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do wycofywania się z rynku tych mniejszych spółek, które obracały energią, do upadku tych spółek, a to jest w dłuższej perspektywie bardzo niekorzystne działanie dla gospodarki.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mówiąc o wzroście cen energii elektrycznej, musimy też mówić o ubóstwie energetycznym. To niestety zagraża coraz większej grupie ludzi, mieszkańców naszego regionu i Polski, ale regionu również, bo nasza energetyka jest energetyką produkującą coraz droższy prąd, w przeciwieństwie do sąsiadów. Ilu mieszkańców ma kłopoty z tym, ażeby dogrzewać swoje mieszkania? Powstaje pytanie, czy nie powinniśmy zastanowić się nad VAT-em związanym właśnie z energią. Czy nie powinniśmy, szczególnie w ciepłownictwie, jeśli np. korzystanie z gazowej energetyki cieplnej jest obarczone 23-procentowym obciążeniem VAT-owym, a to ta energetyka powoduje, że właśnie produkujemy mniej. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę z tym 2050 r. i dlaczego nie decydujemy się jako rząd na to, ażeby 2050 r. był rokiem skutecznej zeroemisyjnej transformacji, zwłaszcza że jako rząd - jest to w polityce energetycznej - mówicie o energetyce atomowej, ale wydaje mi się, że tak jak ze wszystkim, co robicie, jest to trochę fantasmagoria, trochę brak zdecydowania i trochę brak konsekwencji. Jak bowiem możemy poważnie mówić o wybudowaniu dwóch bloków energetyki atomowej w 2033 r., skoro taki np. Flamanville albo Olkiluoto w Finlandii budowane są od kilkunastu lat i ten proces jeszcze jest niezakończony, gdyż napięcie między tzw. generacją III+ a przyszłościową IV i zabezpieczeniem mieszkańców jest tak istotne? Tak więc musimy też odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu tak naprawdę służy pomoc publiczna, bo wydajemy olbrzymie pieniądze na to, ażeby pomóc np. energetyce konwencjonalnej, a zdecydowanie mniejsze pieniądze wydajemy na to, ażeby pomóc energetyce odnawialnej. I teraz jest między tymi dwiema pomocami publicznymi takie napięcie, bo tak naprawdę pieniądze wydawane na to, żeby zabezpieczyć konwencję, służą tylko temu, żeby zakonserwować stary system - i tu wydajemy olbrzymie pieniądze - a wydajemy zdecydowanie małe pieniądze właśnie na OZE, które ma spowodować, że nasza energetyka będzie o wiele tańsza. Rząd musi wreszcie też stanąć w prawdzie i powiedzieć: tak, musimy zrobić sprawiedliwą transformację energetyczną i sięgając po pieniądze europejskie, musimy także jako odpowiedzialny rząd zabezpieczyć regiony typu Bełchatów, typu Konin z Ościsłowem. Musimy też odpowiedzieć na pytanie, czy i jak zrekompensujemy tym regionom to, że przez wiele dziesiątek lat dawały energię Polsce, [[Oklaski]] naszemu krajowi i przyczyniały się do rozwoju, a teraz muszą w jakiś sposób zregenerować się społecznie, żeby zmienić paradygmat rozwoju gospodarczego, ale także ekologicznie, środowiskowo. To są bardzo ważne rzeczy i rząd nie może zamykać oczu i nie odpowiadać na te sprawy.

Mówiliśmy o tym, że dochodziło do spekulacji na Towarowej Giełdzie Energii.

Będzie to powodowało, że my naprawdę będziemy skansenem energetycznym Europy i będziemy skazani w pewnym momencie nie na suwerenność energetyczną (Dzwonek), ale na podległość energetyczną dzięki taniemu prądowi z Niemiec, z Czech i ze Słowacji. Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pana Tadeusza Skobla. Bardzo proszę, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tych pytań było bardzo dużo.

Panie pośle, uprzejmie zapraszam na stronę Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Energii. Te dwa dokumenty tam wiszą.

Tak że nie ma żadnych tajemnic w tym względzie. Te dokumenty są przygotowane i są odpowiednio przedstawione tym organom, którym trzeba. Polityka jeszcze nie.

Tak że od strony społecznej, konsultacyjnej to, co należało zrobić, zostało zrobione.

Myślę, że warto powiedzieć, co on zawiera. Pewne ogólniki ominę, ale przytoczę pewne kluczowe rzeczy.

Wrócę do niej na końcu.

Państwo pytacie: Jaki kierunek? Ten kierunek to jest kierunek OZE. Oczywiście mamy świadomość tego, że OZE nie załatwi nam wszystkiego. OZE potrzebuje źródeł, które by występowały wtedy, kiedy nie wieje i nie świeci. Pewnie przyjdzie taki czas, kiedy trzeba będzie to zrobić.

Pozostałe to biogaz, biomasa i elektrownie wodne.

Tak faktycznie było.

Myślę, że jak państwo czytacie i przeglądacie prasę, również niemieckojęzyczną, i te informacje, które stamtąd płyną, widzicie państwo, że ten problem. Niemcy poszli może troszeczkę za daleko i dzisiaj mają pewien problem, jeżeli chodzi właśnie o tę kwestię. Dzisiaj wszystkie inne kraje również chcą jak gdyby wejść w ten system. Obecny szef Niemiec w zakresie gospodarki energii zaproponował 1000 m odległości od zabudowań.

Wiatraki są bardzo dobre wtedy, kiedy wieje. Ale państwo macie świadomość tego, że w momencie, kiedy mocno wieje, a takie sytuacje były jeszcze w poprzednim roku, w grudniu.

Drodzy Państwo! Ale my dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej i mamy określony poziom wymiany systemowej w Unii. Do tej pory to było 30%, a jesteśmy zobowiązani do tego, by udostępnić swoje moce na przesyle do 70%.

Ta, która jest najtańsza - wchodzi, ta, która jest droższa - nie wchodzi. I choćby ona była najlepsza i nasza, to jest problem. Jest problem, którym na pewno z jednej strony jest bezpieczeństwo.

Z drugiej strony wszyscy państwo dopominacie się o tanią energię. Tania energia musi być elementem kompromisu pomiędzy tym, co się wprowadza w zakresie energetyki odnawialnej. Energetyka odnawialna ma pierwszeństwo w wejściu do systemu energetycznego. To nie jest tak, że ktoś odcina energię odnawialną. Jeden przypadek może być.

Wiem, że pytań jest wiele, przynajmniej w tych systemowych kwestiach chciałem odpowiedzieć. Na lądzie zostały uruchomione wszystkie wiatraki, które miały pozwolenie na budowę, a zasadę 10H spełniają, to poszło.

Mnie osobiście zależało na tym, żeby pokazać społeczeństwu: zobaczcie, macie szansę, możecie w to zainwestować, wejść, spróbować. Weszli. Bardzo dużo osób weszło, jeżeli chodzi o „Mój prąd” cztery pierwsze miesiące - 21 tys. wniosków, kwota 104 mln zł, 117 MW mocy więcej.

Drodzy państwo fotowoltaika nie potrzebuje żadnych pozwoleń na budowę. To się robi szybko. Nam zależało na tym, żeby mechanizm był prosty. Fotowoltaikę się montuje, przedstawia rachunek, zwraca się, w miarę szybko przechodzi to przez ministerstwo wtedy energii, dzisiaj: aktywów, do środowiska do wypłaty i to działa. Zadziałało, na pewno trzeba to wykorzystać. Zależało nam na tym, żeby zachęcić społeczeństwo do korzystania z fotowoltaiki, natomiast musimy mieć świadomość, że fotowoltaika to jest 11,5, 12% z mocy energii, o ile 30, 40% to dobra elektrownia, czy nawet 50, to tutaj tylko 15, 11, 12, czyli mamy - świeci, nie mamy - trzeba wziąć.

Jak jest fotowoltaika, to trzeba zapłacić nie 100% w odbiorze, w relacjach 1 do 1, tylko mniej. Drodzy państwo, system trzeba skompensować.

Czy to jest wystarczające? Spółki sygnalizują, że w niektórych przypadkach nie, że to jest nieco za mało, ale zostawiamy to jeszcze do szczegółowej analizy, dlatego też ilość energii, która może być tłoczona do systemu z fotowoltaiki, z wiatraków, też musi być trzymane w pewnych ryzach. Co się dzieje, gdyby ta energia nagle wtłoczona weszła do systemu? Dzieje się to, że zamiast tej częstotliwości, którą dzisiaj mamy, pojawia nam się inna częstotliwość w sieci.

Jak ma być tyle herców, to może być 1,5% więcej, nieco mniej, ale w odpowiednich granicach. Drodzy państwo, w pewnym momencie Czarnogóra i ten rejon wyłączyły się z systemu, niby prawie nic, wydawało się. W ciągu miesiąca z tytułu częstotliwości, a zegary chodzą na częstotliwość, taktowane są częstotliwością sieci, doszło do ok. 6, 8, 9 minut spóźnienia. Mówię o tym dlatego, że ważną rzeczą jest, by zapewnić nie tylko bezpieczeństwo, ale i odpowiednią jakość energii elektrycznej. Musimy rozwijać energetykę, i powinniśmy, fotowoltaiczną, wiatrową, ale jednocześnie musimy przystosowywać sieci energoelektryczne do odbioru tej energii, przesłania dalej.

Jeżeli cokolwiek jest wyłączone, to to, co jest wyłączone w zakresie związanym, powiedzmy, z koniecznością ograniczenia z takiego względu, że tej mocy jest za dużo. Co się wtedy dzieje? Zobaczcie państwo, z punktu widzenia ekonomicznego, wielu z państwa w tej ekonomice siedzi, jak energia. Jeżeli jest mniejsza produkcja, to jednostkowe koszty wpływające na cenę są większe.

To jest problem społeczny, który musimy rozwiązać. Pod względem ekonomicznym nie jest to może najszczęśliwsze, ale daje szansę na kontynuację.

Jeden i drugi tani nie jest. Tak czy inaczej odpowiem tylko tyle, że jako alternatywną, może nie alternatywną, tylko uzupełniającą w zakresie energetyki jądrowej planujemy również jedną z lokalizacji - badamy w tej chwili ten teren - w rejonie Bełchatowa, sprawdzamy, czy tam blok energetyki jądrowej by się mógł pojawić. Jeżeli tylko warunki geologiczne pozwolą, to będzie to bardzo dobry teren, by tak się stało. Odbiór energii - cały system energetyczny jest przygotowany właśnie do tego.

Ja wiem, właśnie, Wysoka Izbo, przede wszystkim chciałam podkreślić, że przedłużyłam wypowiedź pana ministra na wyraźne życzenie opozycji.

My się zgadzamy z tym, że te problemy trzeba rozwiązać. Przekażemy państwu, w jaki sposób chcemy to zrealizować w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Ta wypowiedź kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 23. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 65) Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Szymona Giżyńskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę, panie ministrze.

projektowanej ustawy w zasadzie uzasadnia do końca intencje, ponieważ kompetencje w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych obecnie podzielone są między Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, czyli IJHARS, która obejmuje produkcję, hurt i kontrolę graniczną, oraz Inspekcję Handlową zajmującą się obrotem detalicznym. Ponieważ jest tak, że są to z oczywistych względów działania komplementarne, do tego inspekcje prowadzą swoją działalność na poziomie i podstawie tych samych przepisów, tej samej ustawy i jednocześnie na tym samym szczeblu - wojewódzkim, no to aż się prosi, żeby w tym procesie scalania inspekcji żywnościowych w Polsce, tak ogólnie to nazywając, poczynić bardzo oczywisty krok. Oczywisty, dlatego że w tych warunkach pozostaje po prostu tylko czynność urzędnicza spajania aktywów i jest to czynność o tyle prosta, że bardzo łatwo nie tyle wydedukować i nie tyle założyć, ile spodziewać się najzupełniej oczywistych, pozytywnych skutków. We wszystkich przygotowawczych pracach nikt nie mógł zakwestionować faktu czy oczywistości, która z tych kalkulacji wynika: że pierwszym efektem będzie znacznie szybsze reagowanie na nieprawidłowości pojawiające się na rynku i tym samym szybsze wycofywanie produktu o niewłaściwej jakości handlowej. Także, co oczywiste w równym stopniu, chodzi o krótszy czas kontroli, czyli postępowania kontrolnego, oraz o wyeliminowanie możliwości sprzecznych interpretacji, które się przecież w sytuacjach rozdzielnej kontroli mogą pojawiać, mimo iż praca polega na analizowaniu i realizowaniu, wdrażaniu w życie tych samych dokumentów, o czym wspomniałem. Jest również oczywistością, że nastąpi pełne, sumujące się połączenie potencjałów ludzkich, ale także rzeczowych i laboratoriów, które będą w to włączone, czyli wszystkich zasobów będących już w tej chwili aktywami jednej inspekcji.

To są informacje dla Wysokiej Izby, które oczywiście mają jedną intencję: prośby o wsparcie, poparcie tej ustawy. Tę prośbę chcę wzmocnić i poprzedzić wskazaniem, iż ten projekt ma wymiar wyłącznie pozytywny. Nie skupia się na przezwyciężaniu trudności, jakichś dysfunkcji, lecz wyłącznie na zarządzaniu komplementarnymi aktywami, które znalazły w tym momencie, w tej koncepcji ujście w jednolitej formule jednej inspekcji. Bardzo proszę o poparcie takiego sposobu myślenia i takiego konkretnego zapisu projektu ustawy, który, jak nam się wydaje, jest całkowicie zgodny z naszymi intencjami, a więc funkcjonalny, praktyczny i skuteczny. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy zabierze głos pan poseł Leszek Galemba, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę o przedstawienie stanowiska klubu. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 65. Projekt dotyczy wprowadzenia zmiany polegającej na powierzeniu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zadań w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu, produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Argumentem, który przemawia za takim rozwiązaniem jest fakt, że nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych jest sprawowany przez IJHARS i Inspekcję Handlową na podstawie tych samych przepisów. Przewiduje się, że stworzenie jednego organu urzędowej kontroli żywności odpowiedzialnego za kontrolę jakości handlowej na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności umożliwi szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości. Rozwiązaniem najkorzystniejszym jest powierzenie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych organowi kontrolnemu podległemu ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, który sprawuje nadzór nad realizacją zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Wobec powyższego uzasadnione jest, aby organ urzędowej kontroli żywności sprawujący nadzór nad jej jakością w produkcji i w obrocie detalicznym podlegał ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych. Z kolei prawidłowe stosowanie materiałów i wyrobów w kontakcie z żywnością może mieć wpływ na jakość handlową oferowanych z użyciem takich wyrobów i materiałów artykułów rolno-spożywczych, dlatego Inspekcja Handlowa weryfikowała stosowanie przez przedsiębiorców wymagań dotyczących materiałów i wyrobów. Projektowane skoncentrowanie w ramach jednej inspekcji odpowiedzialności za kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych pozwoli na szybsze reagowanie i wyjaśnienie wątpliwości związanych ze spełnianiem przez podmioty produkujące i wprowadzające do obrotu wyroby spożywcze. Działanie jednej inspekcji skróci czas niezbędny do zakończenia postepowania kontrolnego oraz wyeliminuje możliwą obecnie ewentualność innej interpretacji przepisów prawnych w związku z wprowadzaniem kontroli przez jedną albo drugą służbę kontrolną. Pozwoli to w założeniu na szybsze wycofanie z rynku produktów nieodpowiadających wymaganiom przepisów prawnych, co przyczyni się w konsekwencji do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstw i ujednolicenia kryteriów oceny. W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości wnoszę o uchwalenie tej ustawy i dalsze nad nią procedowanie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi pan poseł Tomasz Lenz. Zapraszam.

Wysoka Izbo! Dyskutujemy dzisiaj nad projektem dotyczącym kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych. Obecnie kompetencje w zakresie nadzoru nad jakością handlową tych produktów należą do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, nie dotyczy to jednak kwestii obrotu detalicznego. Kontrolą na tym etapie zajmuje się Inspekcja Handlowa. Projekt zakłada powierzenie wszystkich zadań dotyczących kontrolowania jakości tych artykułów jednemu organowi urzędowej kontroli żywności. Uważamy, że jest to dobre rozwiązanie. W modelu, jaki obecnie jest praktykowany w Polsce, nadzór całej drogi, jaką przebywa żywność, od produkcji po jej sprzedaż detaliczną wymaga zaangażowania dwóch instytucji, które różnią się usytuowaniem w strukturach administracji rządowej. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podlega ministrowi rolnictwa, zaś Inspekcja Handlowa - prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taka sytuacja stwarza ryzyko zbyt wolnej reakcji na zagrożenia, jakie pojawiają się dla ekonomicznych i zdrowotnych interesów konsumentów. Proponowane zmiany mają swoje argumenty prawne, gdyż nadzór w obydwu inspekcjach jest wykonywany na podstawie tych samych przepisów, czyli ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Powierzenie kompetencji w zakresie kontroli żywności zarówno w produkcji, jak i w handlu detalicznym jednej instytucji nadzorczej pozwoli efektywniej i z większą korzyścią dla konsumentów, czyli tak naprawdę dla nas wszystkich, działać na rzecz poprawy jakości produktów dostępnych w naszym kraju, umożliwi też szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości, a co za tym idzie - szybsze wycofywanie produktów niespełniających norm jakościowych. Istotne jest także wprowadzenie jednolitych procedur kontrolnych w obszarze jakości handlowej na wszystkich etapach obrotu artykułami rolno-spożywczymi, w tym możliwość stosowania jednolitych wytycznych dla prowadzenia postępowania kontrolnego, wyspecjalizowania laboratoriów i stosowanej metodyki badań, a także efektywniejsze wykorzystywanie inspektorów. To również wpłynie na skuteczność działań inspekcji i ich wyniki. Zmiany, jakie przewiduje ten projekt, będą miały także wpływ na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż dzięki odciążeniu prezesa tego urzędu od spraw związanych z kontrolą żywności w obrocie detalicznym będzie on mógł lepiej skoncentrować się na wykonywaniu innych istotnych kompetencji, które mu przysługują.

W tym gronie są tak ważni producenci żywności, jak: Dania, Francja czy Holandia. Jako klub uważamy, że to rozwiązanie ma szansę sprawdzić się w Polsce.

Chodzi tu o brak określenia, czy w ramach informacji, jakich główny inspektor może zażądać od inspektorów wojewódzkich, mieszczą się dane osobowe. Prawo dotyczące przetwarzania danych osobowych nakazuje zbieranie tylko takich informacji, które są niezbędne ze względu na cel ich gromadzenia. Dlatego przychylamy się do sugestii prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych co do doprecyzowania przepisów w tym zakresie.

Liczymy, że i te kwestie będą uzupełnione w toku prac parlamentarnych. Po uwzględnieniu tych poprawek jako klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej będziemy głosować za przyjęciem niniejszej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu klubu parlamentarnego Lewica w pierwszej kolejności wystąpi pan poseł Marcin Kulasek. Bardzo proszę o przedstawienie stanowiska klubu. W imieniu klubu Lewica pragnę zaprezentować pierwszą część stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Polska żywność jest powodem do dumy. Gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, były to 4 mld. Za tym sukcesem nie nadąża organizacja inspekcji dbających o jakość żywności. Lewica od blisko 10 lat apeluje o utworzenie jednej, zintegrowanej inspekcji. W ostatnim roku o utworzenie jednej inspekcji wnioskował również NIK. W przeciwnym razie do polskich, europejskich konsumentów będą docierać informacje o uboju chorego bydła czy niepokojących, rosnących pozostałościach antybiotyków w polskim mięsie. Proponowana przez resort rolnictwa ustawa to krok niewystarczający, ale krok w dobrą stronę. Dlatego Lewica opowie się za kontynuowaniem prac nad projektem i skierowaniem go do dalszych prac w komisji. Już teraz jednak w Sejmie muszą wybrzmieć ważne kwestie. Po pierwsze, przewidujecie dla Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych znacznie więcej obowiązków, ale tylko niewiele więcej etatów. Po kilka nowych etatów na województwo to zdecydowanie za mało. Kontrola żywności nie będzie skuteczna, kiedy pracownicy inspekcji będą zarabiać trochę powyżej płacy minimalnej. W ten sposób nigdy nie stworzymy sprawnego systemu kontroli. Po trzecie, w projekcie nie ma listy laboratoriów, które przejdą wraz z kompetencjami do IJHARS. Po czwarte, należy wrócić do dyskusji na temat wyłączenia IJHARS z administracji zespolonej. Sytuacja, w której inspekcje wojewódzkie podlegają wojewodom, powoduje rozproszenie zasobów i zmniejszenie skuteczności kontroli. Ustawa zwiększa rolę głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, co należy ocenić pozytywnie. Ta zmiana jest jednak niewystarczająca. Po piąte, w uzasadnieniu ustawy na str. 10 czytamy, że inspekcja handlowa nie posiada baz danych, które służyłyby analizie prawdopodobieństwa naruszenia praw w zakresie bezpieczeństwa żywności. W oparciu o jakie dane troszczycie się o bezpieczeństwo Polek i Polaków? Polacy mają prawo mieć pewność, że żywność, którą mają na talerzu, jest bezpieczna. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przedłożony projekt budzi istotne zastrzeżenia dotyczące kompetencji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Chodzi o obowiązek prowadzenia kontroli prawidłowości dokonywanych transakcji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Gwarancji, realizowanych w ramach wspólnej polityki rolnej. Trzeba podkreślić, że kontrole takie nie mają nic wspólnego z problematyką jakości żywności, dotyczą tylko problematyki sposobu wydatkowania środków publicznych w ramach wspólnej polityki rolnej. Tego rodzaju kontrole powinny być prowadzone przez stosowne, wyspecjalizowane krajowe agencje płatnicze, takie chociażby jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Problem ten jest istotny także z dwóch innych powodów. Po pierwsze, inspektorzy zatrudniani w strukturach Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych to przede wszystkim fachowcy o kompetencjach w kwestiach jakości żywności, a nie w kwestiach finansów i rozliczeń transakcyjnych. Po drugie, rozszerzenie nadzoru o szczebel handlu detalicznego przysporzy inspektorom znacznie więcej kontroli, a więc będzie od nich wymagać znacznie większego zaangażowania czasowego, co może w sposób istotny ograniczyć skuteczność nadzoru o charakterze finansowo-rozliczeniowym. Podsumowując, proponowane zwiększenie uprawnień Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, szczególnie w zakresie skarbowo-podatkowym, wpisuje się w niepokojący i coraz bardziej powszechny trend zwiększania siły instytucji kontrolujących kosztem przedsiębiorców. Stąd też wnosimy o skierowanie omawianego projektu do pracy w komisjach. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Kukiz15 głos zabierze pan poseł Jarosław Sachajko. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! W imieniu klubu Koalicji Polskiej mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Tu krótko można powiedzieć, że ta ustawa idzie w dobrym kierunku. Wszyscy się zgadzają, że powinna być przyjęta, tylko czy to na pewno jest ta ustawa, którą Prawo i Sprawiedliwość obiecało Polakom. Pod koniec 2017 r. rząd przyjął projekt ustawy o utworzeniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Jest to druk z ubiegłej kadencji, nr 1685. Z jakiegoś powodu Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z tego projektu, nie dotrzymało obietnicy. To już nie pierwszy raz, bo w 2007 r. podobny projekt również Prawo i Sprawiedliwość przygotowało, obiecując Polakom, że będą mieli pewność obrotu żywnością i jakości żywności, i też go nie przyjęło.

Tu państwo wielokrotnie mówili, jakie to jest ważne, wprost było powiedziane, że powołanie nowej inspekcji miało zapewnić efektywne kontrolowanie żywności od pola do stołu, wyeliminowanie przypadków dublowania się i nakładania kompetencji, a także miało obniżyć koszty takiej działalności. Nie potrafią państwo dogadać się w ramach rządu, bo Ministerstwo Zdrowia nie chce oddać trochę kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Co jeszcze mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości? Że połączenie inspekcji odpowiadających za bezpieczeństwo żywności jest jednym ze sztandarowych projektów Prawa i Sprawiedliwości. To co z tym sztandarowym projektem się stało, że on nie jest przyjęty, tylko robią państwo kolejną atrapę, łącząc kawałek inspekcji? Uważam właściwie, że słusznie odbierają państwo kompetencje inspektorowi ochrony konkurencji, prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo to nie działało.

Że będzie to kontrolował. Ostatnia rzecz, jaką muszę powiedzieć, dotyczy niedofinansowania rolnictwa.

A jaka była obietnica Prawa i Sprawiedliwości z 2015 r., kiedy to Prawo i Sprawiedliwość bardzo chętnie krytykowało Platformę Obywatelską i PSL, że za mało finansują? A ile mamy? Gdzie jest spełnianie obietnic co do prawidłowego finansowania rolnictwa, co do przyjęcia ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności? Na to potrzebne są pieniądze, a pieniędzy w budżecie, jak widzimy, nie ma, bo ta zwyżka na tę inspekcję jest minimalna. Dziękuję bardzo. Do pytań zapisało się dwoje parlamentarzystów. Zamykam listę. Wyznaczam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Porządkuje on kwestie związane z odpowiedzialnością za jakość handlową artykułów rolno-spożywczych i, przede wszystkim, służy bezpieczeństwu konsumenta. To jest, myślę, najistotniejsze, najważniejsze. W związku z tym mam pytanie: Jak wnioskodawca widzi dalszą rolę Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w tym wielkim systemie nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi? Czy wnioskodawca dostrzega potrzebę dalszego wzmacniania tej inspekcji i od strony merytorycznej, i od strony etatowej? Dziękuję bardzo. I zapraszam panią poseł Annę Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Z mojej strony - i myślę, że ze strony wszystkich producentów, przedsiębiorców - wielkie ukłony i wielkie podziękowania za tę ustawę.

Nikt nie lubi być kontrolowany, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo żywieniowe, bezpieczeństwo żywności wymaga, aby takie kontrole się odbywały. Przedsiębiorcy też to rozumieją. A więc bardzo się cieszę. Mam natomiast pytanie: Czy ta nowa inspekcja będzie miała kompetencje do kontroli na wszystkich etapach, czyli od momentu produkcji do etapu wytworzenia i wprowadzenia do obrotu danego produktu żywnościowego?

Zapraszam, panie ministrze.

Wysoki Sejmie!

Chcę odpowiedzieć panu posłowi Marcinowi Kulaskowi z Lewicy, że lista laboratoriów jest dołączona do oceny skutków regulacji i obejmuje pięć laboratoriów: w Katowicach, w Kielcach, w Olsztynie, w Poznaniu i w Warszawie.

Po pierwsze, pozostawienie administracji zespolonej w układzie zależności od wojewodów ma swoje uzasadnienie i wielokrotnie na ten temat mówiliśmy.

To może zrobić tylko centrum, może to zrobić główny inspektor i myślę, że to wszystko jest komplementarnie ustawione. Takie jest założenie.

Otóż jeden z mówców jako jedyny w zasadzie wykorzystał ten projekt do tego, żeby powrócić do pewnych motywów czysto politycznych, przerzucających dyskusję na zupełnie inne tereny. Przypominało mi to wczorajszą dyskusję dotyczącą ustawy o ASF.

Na tym polega polityczna wolność i konieczność niczym nieskrępowanej dyskusji politycznej - ale w obrębie zaproponowanego tematu.

Szanowni państwo, jest tak, że zarówno ustawa weterynaryjna - która też niebawem, mam nadzieję, będzie absorbować Wysoką Izbę, bo już jest na tyle przygotowana, że za kilka tygodni będzie także przedmiotem naszych prac w Sejmie - jak i ta dzisiejsza ustawa są dokładnie krokiem w tym kierunku. Tam to, co się da scalić, bez polemik, bez jakichkolwiek kontrowersji.

Przewidujemy to, dofinansowujemy.

To jest założenie ustawy weterynaryjnej, o której dzisiaj nie mówimy, więc na tym kończę. To, co się da szybko skorelować, połączyć, to robimy. Przecież nie było żadnych merytorycznych kontrowersji w odniesieniu do tego pomysłu, co bardzo, ogromnie cieszy.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 65, do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 3. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? W związku z tym listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam za zamkniętą. Głos jako pierwszy zabierze pan poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Chciałbym w swym oświadczeniu poruszyć kwestię obwodnicy dla miasta Kalisza, które jako miasto tej wielkości jest ewenementem w skali kraju, gdyż takowej obwodnicy nie posiada. Obwodnica Kalisza to ważna inwestycja, o której budowę czynię starania od momentu, kiedy zostałem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania z prezydentem miasta Kalisza, które miało miejsce w kwietniu 2019 r., zdecydowana większość parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości zaakceptowała tzw. trzeci wariant budowy obwodnicy. Jedno z najważniejszych kryteriów, które brane są pod uwagę, dotyczy wielkości natężenia ruchu. W Kaliszu badania takie prowadzi od 2016 r. miejski zarząd dróg i komunikacji. W tym miejscu pojawia się pytanie: Dlaczego takich badań nie prowadziły władze miasta Kalisza za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL? Wówczas, kiedy prezydentem miasta Kalisza był obecny senator Platformy Obywatelskiej pan Janusz Pęcherz, a funkcję wiceprezydenta pełnił jeden z prominentnych działaczy Platformy Obywatelskiej pan Dariusz Grodziński. Dlaczego nie wykorzystano tego czasu, kiedy większość w Radzie Miejskiej Kalisza, w Sejmie i w Senacie miała koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego? Bez wątpienia brak takich pomiarów opóźnił w znaczący sposób realizację tej jakże potrzebnej dla miasta Kalisza inwestycji. Korzystając z okazji, muszę także wskazać polityczne nieróbstwo w omawianej kwestii moich poprzedników, parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy nie potrafili doprowadzić do tego, aby wpisać do „Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023” budowę obwodnicy Kalisza.

W tym miejscu pragnę podkreślić, że wiele miast w Polsce zyskało obwodnicę przy znacznie mniejszym natężeniu ruchu pojazdów. Równie dużo pojazdów, w tym wiele ciężarówek, przemieszcza się przez Kalisz na osi wschód - zachód od strony Łodzi i Sieradza oraz Leszna i Poznania. Podczas rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wiele razy władze miasta Kalisza i posłowie Prawa i Sprawiedliwości z okręgu kalisko-leszczyńskiego zwracali uwagę na ten problem, czyli wyrzucenie, w cudzysłowie oczywiście, tranzytu poza miasto na osi drogi krajowej nr 12.

Mam wielką nadzieję, że budowa obwodnicy dla miasta Kalisza, która to inwestycja pozwoli odciążyć miasto od transportu samochodowego, stanie się w niedługiej perspektywie realna. Budująca jest też informacja, że obecnie analizowane są różne możliwe inwestycje, jakie mogą zostać zrealizowane, wraz z potencjalnym harmonogramem realizacji, jak i to, że zadanie dotyczące budowy obwodnicy Kalisza jest rozważane w ramach tegoż programu. Równie budujące jest to, że prawie wszyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości w Wielkopolsce dostrzegają problem braku obwodnicy miasta Kalisza i rozumieją pilną potrzebę wpisania tej inwestycji właśnie w ten program budowy 100 obwodnic dla miast w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie jest dostępna w Systemie Informacyjnym Sejmu. Na tym kończymy 3. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.